Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi szereg programów, które mają na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Tych programów naprawdę jest dużo i środki, które rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznacza na te programy, są znacząco większe niż w poprzednich latach. Przypomnę tylko, że w roku 2015 była to kwota ok. 15 mld.

Przypomnę - obok szczegółowego pytania, które chcę zadać, dotyczącego opieki wytchnieniowej i tego programu - że jest również bardzo duży program „Dostępność+”, są programy dedykowane osobom starszym, seniorom, są programy wsparcia dla środowisk, organizacji pozarządowych, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej, ZAZ-y, tak że tych programów jest bardzo dużo.

Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. O udzielenie odpowiedzi proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pana ministra Pawła Wdówika. Bardzo proszę, panie ministrze.

Wysoka Izbo! We wrześniu br. zakończył się nabór wniosków związanych z przekazaniem rządowych środków finansowych na opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób starszych i niesamodzielnych.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Program jest realizowany w trzech formach. Pierwsza forma to jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego. To się może odbywać w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia albo w innym miejscu wskazanym przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię realizatora programu, czyli można wskazać nawet dom sąsiada, ale pod warunkiem że on spełnia kryteria, których spełniania wymagamy od miejsca zapewniającego odpowiedni standard i dostępność dla osoby z konkretną niepełnosprawnością. Druga forma to świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Ostatnią formą jest inne miejsce wskazane przez uczestnika programu, z tym że też musi zostać zaakceptowane przez organizację realizującą ten program. I trzecia forma: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa, w tym psychologicznego, lub terapii oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. W ramach programu ustala się następujące limity: limit 240 godzin w przypadku opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, limit 14 dni w przypadku opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego i limit 20 godzin w przypadku opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa. Jeżeli chodzi o to, jakie mamy oferty, 115 uprawnionych podmiotów, tj. organizacji pozarządowych posiadających statut, w którym jest zapisana działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością, oraz prowadzących działalność na rzecz dzieci z niepełnosprawnością, złożyło 157 ofert, w tym 43 oferty na rok 2020 i 114 ofert na rok 2021. Zgodnie ze złożonymi ofertami ogółem planowana liczba uczestników programu to ponad 7200 osób. 72% z nich stanowią osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a 28% stanowią dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Uprawnione podmioty przesyłały swoje oferty konkursowe w terminie do 16 października. Przedłużyliśmy ten termin, bo początkowo było ich mało. Dodatkowo chcę jeszcze zwrócić uwagę, że na realizację usług opieki wytchnieniowej za pośrednictwem i z udziałem samorządów, gmin i powiatów w zeszłym roku przeznaczyliśmy 110 mln zł, z czego przekazano 23 mln.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze.

Pani poseł, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Program na lata 2020-2021 „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” po raz pierwszy skierowany jest także do organizacji pozarządowych posiadających statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz takich, które prowadzą taką działalność przez okres co najmniej 3 lat od dnia złożenia oferty. Czy mógłby pan odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu przeznaczone na ten program środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę. Szanowna Pani Poseł! Szanowni Państwo! Ten program w całości jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, czyli te wszystkie kwoty, o których mówiłem, które są przekazywane do samorządów czy do organizacji, są środkami Funduszu Solidarnościowego.

Zobaczymy, jak będzie wyglądała realna kwota wykorzystana, natomiast wydaje się, że te 30 mln w całości nie zostanie skonsumowane. I na przyszły rok przewidzieliśmy po 50 mln dla samorządów i organizacji pozarządowych, z tą różnicą, że tu jesteśmy już gotowi pokrywać do 100% kosztów. Ważną rzeczą jest, bo to może potem być istotny aspekt analizy dla niektórych z państwa, że 100% wniosków samorządów zostało zrealizowanych. Każdy, kto chciał dostać, dostał pieniądze. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie w sprawie nierozliczenia umowy na zakup respiratorów oraz braku celowości, gospodarności i transparentności przy dokonywaniu zakupów związanych z COVID-19 - skierowane do ministra zdrowia. Pytanie przygotowane przez posłów Michała Szczerbę i Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym przede wszystkim pokłonić się polskim kobietom, polskim dziewczynom, które dzisiaj uczestniczą w całym kraju w Ogólnopolskim Strajku Kobiet. Każdego dnia budzicie się z pewną niepewnością, z lękiem o życie, o zdrowie swoich najbliższych, z pytaniami, czy pojawi się koronawirus, czy wtedy, kiedy się pojawi, zostanie udzielona osobie najbliższej pomoc, znajdzie się miejsce w szpitalu, znajdzie się respirator. Wczoraj mieliśmy podane dane: zajętych 1078 respiratorów na 1594 przygotowanych. Ale, szanowni państwo, te dane trzeba również rozważać w kontekście umów, które zawierało Ministerstwa Zdrowia, umów, z których wyszło niewiele, a tak naprawdę - bardzo niewiele. Do tej pory, szanowni państwo, z umowy zawartej przez ministra Szumowskiego 14 kwietnia nie dostarczono 1041 respiratorów. 1041 respiratorów to jest mniej więcej tyle, ile w tej chwili respiratorów jest zajętych. Ale co najważniejsze, mamy do czynienia z przykładem naprawdę niebywałej niegospodarności, niecelowości, ale również działań, które zawstydzają i powinny zawstydzać Ministerstwo Zdrowia. Do tej pory handlarz bronią, który był kontrahentem Łukasza Szumowskiego, nie zwrócił blisko 70 mln zł. Przez pół roku Ministerstwo Zdrowia występuje jak taka kasa pożyczkowa, która pozwala zasilać start-up, który następnie obraca pieniędzmi ministerialnymi - nie wiadomo gdzie, nie wiadomo, w jakim celu. Pani Minister! Jak wygląda rozliczenie z handlarzem bronią? Kiedy te pieniądze zostaną zwrócone? Czy powiadomiliście prokuraturę, CBA, czy skierowaliście sprawę do sądu? Czy macie świadomość tego, że nie podejmując tych działań, również narażacie się na odpowiedzialność karną? Odpowiedzi na pytanie udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pani minister Józefa Szczurek-Żelazko. Bardzo proszę, pani minister. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pandemia była i jest zjawiskiem, które postawiło ogromne wyzwania przed rządami nie tylko Polski, ale wielu różnych krajów Europy i świata. Przed pierwszymi przypadkami, które pojawiły się w Polsce, jak wielokrotnie pan minister Szumowski i pan minister Niedzielski państwa informowali, dokonywaliśmy szczegółowych analiz zasobów, które są w systemie ochrony zdrowia, jak również dokonywaliśmy szczegółowych analiz płynących z różnych krajów, a świadczących o przebiegu epidemii. Z naszych analiz wynikało, że te zasoby, jeżeli chodzi o potencjał łóżkowy, wyposażenie łóżek czy też wyposażenie stanowisk do intensywnej terapii, powinny odpowiadać na potrzeby Polaków. Ale patrząc na to, co się dzieje we Włoszech, co się dzieje w Hiszpanii. Mieliśmy świadomość, że taka sytuacja może pojawić się również w Polsce.

Dlatego też 14 kwietnia 2020 r. została zawarta przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra zdrowia umowa ramowa z firmą E&K sp. z o.o., której przedmiotem było ustalenie warunków współpracy dotyczącej zakupów dokonywanych przez Ministerstwo Zdrowia i dostaw dokonywanych przez tę firmę. Zgodnie z brzmieniem §1 tejże umowy ramowej w dniu 14 kwietnia Skarb Państwa reprezentowany przez ministra zdrowia zaakceptował ofertę tej firmy i podpisał zamówienie na dostawę 1241 respiratorów. Dostawa respiratorów miała być zrealizowana w kilku etapach.

Przedmiotem zamówienia były respiratory, tak jak powiedziałam, które miały służyć pacjentom w stanie zagrożenia życia. Były to respiratory różnych typów, różnych modeli, ale oczywiście te respiratory, zgodnie z tą podpisaną umową, miały mieć wszelkie certyfikaty i spełniać wszelkie warunki, które są określone w przepisach zarówno międzynarodowych - tutaj odnoszę się do przepisów unijnych - jak i w naszych przepisach krajowych. W związku z tym zamówiono cztery rodzaje respiratorów. Pierwszy to były respiratory w ilości 200 sztuk, które miały trafić do Polski w kwietniu - w ilości 25 sztuk, w maju - co najmniej 50 sztuk, następnie w czerwcu - pozostałe 125 sztuk.

W przypadku tych respiratorów została dokonana przedpłata w 100%. Kolejny rodzaj respiratorów, który objęty był tą umową, to była ilość 196 sztuk i również realizacja tej umowy miała być etapami: w maju - 46 sztuk, w czerwcu - 150 sztuk.

Dokonano przedpłaty w wysokości 65%, a 35% po dostawie każdej partii. Kolejne respiratory w ilości 200 sztuk, następnie 645 sztuk (Dzwonek) miały być przekazane do końca kwietnia i do końca czerwca i również były objęte przedpłatami. W trakcie realizacji umowy ta spółka nie wywiązała się z terminów dostaw, a tym samym Skarb Państwa odstąpił od poszczególnych części umowy wykonawczej. Ostatecznie firma dostarczyła 200 respiratorów, to jest 50 sztuk respiratorów firmy Draeger, jedna sztuka po 45 tys. euro, i 150 respiratorów, jedna sztuka po 44 700 euro.

W związku z ww. odstąpieniami, zgodnie z postanowieniami umowy ramowej, naliczone zostały również kary umowne oraz wysłane wezwania do zapłaty kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku opóźnienia w zapłacie.

z pismem przekazanym przez firmę 14 sierpnia spółka zobowiązuje się do zwrotu naliczonych zaliczek w terminie do 30 października tego roku.

Dziękuję bardzo, pani minister. Z pytaniem uzupełniającym pan poseł Dariusz Joński. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Pani Minister! Ja powiem dokładnie: 73 966 tys. zł, tyle brakuje. Kiedy z panem posłem Szczerbą nagłaśnialiśmy tę sprawę w maju i czerwcu, pan premier Morawiecki mówił: Nie słuchajcie brzęczących much. Szumowski mówił: Nie ma mowy o oszustwie, pieniądze wrócą, respiratorów nie zabraknie. Przyczyna: brakuje respiratora. Chwilę później w szpitalu bielańskim w Toruniu właśnie to się dzieje. Państwo podejmujecie decyzję, aby zwiększyć tę ilość. Na dzisiaj starczy tych respiratorów na 7 dni. My słyszymy, że za tym wszystkim stoi Agencja Wywiadu, pani minister. Zysk z operacji miał być przekazany na fundusz operacyjny. Operacja się udała, tylko pacjent zmarł. To jest największa afera w historii Ministerstwa Zdrowia. Pieniądze powinny zostać zwrócone. A jeśli nie mają, to niech pracują na oddziałach Dziękuję. Pani minister, bardzo proszę. Proszę o udzielenie odpowiedzi.

Szanowni Państwo! Te respiratory, które zostały dostarczone przez tę firmę, ale nie tylko przez nią, bo równocześnie zostały zakupione i przekazane do Agencji Rezerw Materiałowych respiratory z innych firm, są na bieżąco przekazywane do podmiotów leczniczych. Jeżeli są takie zgłoszenia, minister zdrowia wydaje dyspozycję i ten sprzęt jest natychmiast wydawany. Chciałabym podkreślić jeszcze jedno: że wojewodowie, analizując sytuację epidemiologiczną na swoim terenie, praktycznie codziennie czy nawet kilka razy dziennie podejmują decyzje o zwiększeniu liczby łóżek przeznaczonych dla tych pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji, ale również dla tych, którzy wymagają leczenia w warunkach intensywnej terapii, czyli chodzi także o zwiększenie liczby łóżek wyposażonych w respiratory. Pamiętajmy, że w naszym kraju mamy ok. 10 tys. łóżek, które są wyposażone w standard obejmujący m.in. respiratory. To są łóżka, które w normalnym trybie funkcjonują w naszych szpitalach.

Tak jak powiedziałam, te dostawy na bieżąco są realizowane, agencja przekazuje respiratory. Reagujemy na każdą potrzebę, również na takie, które panowie posłowie zgłaszają, ponieważ jesteśmy w ciągłym kontakcie. Odpowiadamy państwu na konkretne pytania. Te informacje, które państwo nam przekazujecie, są weryfikowane i natychmiast działania podejmowane są tak, aby pacjenci, którzy potrzebują specjalistycznego sprzętu, potrzebują specjalistycznej opieki, mogli na taką opiekę liczyć. Dziękuję bardzo, pani minister. Przechodzimy do kolejnego pytania, również skierowanego do ministra zdrowia. To pytanie w sprawie wycofywania się szpitali z badań prenatalnych i terminacji ciąż z przyczyn embriopatologicznych. Pytanie zostało przygotowane przez klub Lewica, posłów Krzysztofa Gawkowskiego, Anitę Kucharską-Dziedzic, Jana Szopińskiego, Karolinę Pawliczak, Beatę Maciejewską, Agnieszkę Dziemianiowcz-Bąk, Anitę Sowińską i Zdzisława Wolskiego. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Kilka dni temu społeczeństwo dowiedziało się o skandalicznym postępowaniu dyrekcji Szpitala Bielańskiego, która - zanim orzeczenie quasi-Trybunału Konstytucyjnego zostało opublikowane - wykorzystała je jako pretekst do złamania konstytucyjnego prawa do równego dostępu do ochrony zdrowia i świadczeń gwarantowanych polskim prawem. Powstał okólnik nakazujący odmawianie kobietom terminacji ciąży z przyczyn embriopatologicznych. Dzięki interwencji posłanki Lewicy Wandy Nowickiej Szpital Bielański wycofał się z tej decyzji wskazującej na niedopuszczalną nadgorliwość i lekceważenie litery prawa. W ilu polskich szpitalach mających oddziały ginekologiczno-położnicze wykonuje się pełen pakiet badań prenatalnych i terminację ciąż z przyczyn embriopatologicznych? Ile szpitali odmawia przeprowadzenia procedur medycznych czy badań prenatalnych i terminacji ciąż z przyczyn embriopatologicznych i z wykorzystaniem jakich pretekstów: orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, braku lekarzy, którzy w publicznych placówkach nie kierują się przekonaniami religijnymi, ale stosują się do obowiązującego jeszcze świeckiego państwa i praw pacjenta, obstrukcji czasowej, czyli takiego przedłużania procesu diagnostyczno-decyzyjnego, by legalna terminacja była już niemożliwa? Tu wystarczy przejrzeć odmowy szpitali. Co Ministerstwo Zdrowia zrobiło, jakie wdrożyło procedury dyscyplinujące, by zapewnić wszystkim pacjentkom równy dostęp do świadczeń medycznych gwarantowany prawem? O odpowiedź oczywiście proszę także na piśmie, bo jakoś dziwnym trafem, kiedy zadaję podobne pytania o kwestie łamania praw obywatelskich przez instytucje publiczne kierujące się niepublicznymi przekonaniami kierownictw, nie dostaję miarodajnych odpowiedzi. Dziękuję, pani poseł. Proszę o udzielenie odpowiedzi sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia panią minister Józefę Szczurek-Żelazko. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Myślę, że dla każdego z nas jest to oczywiste, że życie jest najważniejsze: życie dziecka, życie osoby dorosłej, życie seniora. Dlatego działania obecnego rządu, ale również Ministerstwa Zdrowia, realizowane głównie przez ministra zdrowia, zmierzają do zapewnienia tego konstytucyjnego prawa. Pani poseł wspomniała o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który podważył zgodność z konstytucją jednej z trzech przesłanek, które w obecnym stanie prawnym funkcjonowały jako przesłanki umożliwiające terminację ciąży.

Takie przesłanki, te dwie przesłanki zostały. Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się na temat tych dwóch przesłanek. Szanowni Państwo! Jak wszyscy wiemy, bo jesteśmy parlamentarzystami, prawo obowiązuje od momentu opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym, o tej godzinie, mamy taki stan prawny, jaki obowiązywał przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Po sygnałach, o których pani poseł mówi, które pojawiają się w pojedynczych szpitalach, podejmowaliśmy interwencje.

Na dzień dzisiejszy w Ministerstwie Zdrowia nie mamy sygnałów, który szpital odmawia wykonania tychże zabiegów. Szanowni Państwo!

W ostatnim roku, w 2019 r., który jest przedmiotem sprawozdania przyjmowanego przez Sejm, wynika, że w kraju zostały wykonane 174 przypadki aborcji z przesłanek medycznych, które wskazywały na bardzo duże prawdopodobieństwo ciężkiego uszkodzenia płodu.

Szanowni Państwo! Po przeanalizowaniu tych sprawozdań, które do nas wpływają ze szpitali, a w całym kraju, w praktycznie każdym województwie sprawozdawane są te procedury do Narodowego Funduszu Zdrowia, wynika, że większość tych zabiegów jest wykonywana z powodu trisomii, chromosomu 21 i w podziale ze współistniejącymi wadami bądź też bez współistniejących wad. Łącznie ponad 430 zabiegów zostało wykonanych właśnie z tych przesłanek. Oczywiście dużą grupę tych zabiegów stanowią też zabiegi wykonane z powodu mnogich wad płodu, które nie dają szans na samodzielne życie. Wspomniała pani poseł o badaniach prenatalnych. Szanowni państwo, badania prenatalne są prowadzone w Polsce od 2013 r. na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia w zakresie programów zdrowotnych.

Na ten cel z roku na rok przeznaczamy coraz większą kwotę. Jest to też bardzo istotne z punktu widzenia działań naprawczych, które w naszym kraju są wykonywane. Chcę powiedzieć, że jest to. Bo już czas minął, przepraszam najmocniej. Z pytaniem dodatkowym pani poseł Beata Maciejewska, klub Lewica.

Wysoka Izbo! Chciałabym dopytać o jeszcze jedną rzecz. W orzeczeniu pseudo - Trybunału Konstytucyjnego nie ma odniesienia do przerywania ciąży z przyczyn kryminalnych, tzn. wtedy, kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu albo kazirodztwa. Jednak z doniesień medialnych wynika, że właśnie tego. Ma on zmierzać do delegalizacji przerywania ciąży u kobiet pokrzywdzonych przestępstwem gwałtu i kazirodztwa. Chciałabym się dowiedzieć, w ilu polskich szpitalach odmawia się przeprowadzenia procedury terminacji ciąży pacjentkom, które zaszły w nią w wyniku przemocy lub przestępstwa. W ilu się nie odmawia, ale stosuje się obstrukcję czasową? Oczywiście pytam także o to, co Ministerstwo Zdrowia zrobiło (Dzwonek), żeby zapobiec takiemu łamaniu prawa. Jakie ministerstwo planuje wdrożyć procedury, żeby zabezpieczyć prawa pacjentek ofiar przestępstw seksualnych w przypadku analogicznego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego? Bardzo proszę, pani minister. Szanowna pani poseł, jeżeli chodzi o te pozostałe przesłanki, które są zdefiniowane aktualnie w ustawie, to ja podawałam te informacje, że z przyczyn właśnie między innymi. Jeżeli chodzi o ilość dokonanych aborcji w przypadku, gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, w tym roku dokonano trzy takie zabiegi. W kolejnych latach zdarzały się po jednym.

Więc jeżeli istnieją przesłanki ustawowe, takie zabiegi są wykonywane. Tak jak państwu powiedziałam na początku, ze sprawozdań, które są kierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia przez szpitale, wynika, że nie ma na terenie kraju województwa, które nie sprawozdałoby tego typu zabiegów w ostatnich kilku latach. Tutaj również należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty lekarz ma prawo do zastosowania tzw. klauzuli sumienia. Jeżeli wykonanie tego zabiegu jest niezgodne z jego przekonaniami, z jego sumieniem, ma prawo do odmowy. Ale to nie oznacza, że pacjentka pozostaje sama. W tym przypadku podmiot leczniczy czy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wskazuje, gdzie tego typu świadczenie może być wykonywane. Jeszcze chciałabym wrócić do tych badań prenatalnych, bo to jest bardzo istotne, że nie dość, że zwiększamy ilość tych badań, zwiększamy finansowanie, to w Polsce w pięciu szpitalach są również wykonywane zabiegi wewnątrz życia płodowego, które ratują życie, które potrafią niwelować wiele wad i powodować, że dzieci, które po takim zabiegu przychodzą na świat, mają pełne szanse na dobry rozwój i przyszłość. Przekazaliśmy szpitalom ponad 3 mln zł i katalog tych szpitali się rozszerza. Wykonywane są skomplikowane zabiegi np. kardiologiczne, np. zabiegi przy stwierdzeniu przepukliny mózgowo-rdzeniowej, wiele różnych zabiegów, których wykonanie w życiu płodowym albo zmniejszy negatywny wpływ tej wady na przyszłą kondycję zdrowotną dziecka, albo spowoduje, że to dziecko urodzi się całkowicie zdrowe. Dlatego nie zamierzamy ograniczać badań prenatalnych, a wręcz odwrotnie, tak jak pan premier Mateusz Morawiecki wczoraj powiedział, będziemy planować (Dzwonek) rozszerzenie badań prenatalnych, aby wspierać rodziny, wspierać matki w sytuacjach, kiedy dotykają ich tak trudne sytuacje życiowe. Dziękuję. Dziękuję, pani minister. Przechodzimy do kolejnego pytania.

Pytanie zada pan poseł Stanisław Żuk.

Pani Minister! Wysoka Izbo! W Polsce żyje ok. 1 mln osób, u których zdiagnozowano lub wyleczono nowotwór, a prognozy przewidują, że liczba pacjentów onkologicznych może wzrosnąć w ciągu 10 lat o 28%. Z pięciu obszarów działania Narodowej Strategii Onkologicznej najważniejsze z punktu widzenia pacjentów to: dostęp do innowacyjnych terapii, zapewnienie najwyższej jakości standardów diagnostyki i leczenia, zwiększenie dostępu do nowoczesnej aparatury medycznej, prawo do życia bez bólu dla pacjentów onkologicznych. Pacjenci postrzegają polski system opieki onkologicznej jako nieprzyjazny i niewystarczająco skupiony wokół ich potrzeb. Jednym z ważniejszych celów powinno być wprowadzenie nowych procedur zabiegowych, w tym mało inwazyjnych sposobów dawkowania promieniowania medycznego. Ośrodki i podmioty medyczne mające takie możliwości powinny być promowane, a pacjenci muszą mieć zapewniony dostęp do tych innowacyjnych terapii. Rocznie z powodu nowotworów umiera ok. 100 tys. Polaków. Dlaczego więc nie ogłasza się pandemii chorób nowotworowych? Epidemia COVID-19 doprowadziła do sytuacji, w której liczba zgonów wśród chorych onkologicznie będzie rosła bardziej.

Zwracam pani uwagę, że to było niestosowne. Na podstawie art. 175 ust. 2a regulaminu Sejmu stwierdzam, że swoim zachowaniem na sali posiedzeń naruszyła pani powagę Sejmu. Skieruję również tę sprawę do komisji etyki i sprawdzimy, co to jest za numer telefonu. Pani poseł doskonale wie. Pani marszałek, nie ma problemu. Epidemia COVID-19 doprowadziła do sytuacji, w której liczba zgonów wśród chorych onkologicznie będzie rosła bardziej, niż przewidują to prognozy umieralności. Składają się na to: lęk przed COVID-19 opóźniający podjęcie właściwego leczenia, zawieszenie terapii onkologicznych, czasowe zamknięcie oddziałów i szpitali z powodu kwarantanny, przekładanie wielu planowanych zabiegów. Żyjemy w sytuacji nadzwyczajnej. Konieczne jest wykorzystanie potencjału podmiotów medycznych (Dzwonek), które z różnych względów nie świadczą usług medycznych w zakresie diagnozowania i leczenia chorych na raka. Podmioty te powinny zapewnić realizację działań zaplanowanych w Narodowej Strategii Onkologicznej. W związku z tym mam pytania: Ile jest w Polsce niewykorzystanych obiektów mogących świadczyć usługi leczenia chorób nowotworowych w celu zwiększenia dostępu do najnowocześniejszej aparatury medycznej? Dlaczego Narodowy Fundusz Zdrowia nie zawiera kontraktów onkologicznych z SP ZOZ, które posiadają umowę z niezależnym podmiotem gospodarczym na wykorzystanie istniejących i doskonale wyposażonych obiektów związanych z diagnostyką i leczeniem? Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję, panie pośle. Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pani minister Józefa Szczurek-Żelazko. Bardzo proszę, pani minister. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo jest to też okazja, żeby przypomnieć nam wszystkim, przede wszystkim naszym rodakom, którzy słuchają przebiegu obrad, jak ważne są kwestie związane z dbałością o zdrowie, profilaktyką ogólnie rozumianą, ale również profilaktyką onkologiczną, jak przypadek, o którym mówimy. W związku z tym, że rzeczywiście w Polsce zapadalność na choroby nowotworowe bardzo szybko rośnie, mało tego, mamy wskaźniki, które bardzo nas niepokoją, a świadczą o tym, że przeżywalność powyżej 5 lat osób, które doświadczyły choroby nowotworowej, jest znacznie niższa niż w innych krajach Unii Europejskiej, niezbędne było opracowanie konkretnego dokumentu, planu, strategii, która w sposób systemowy, wielosektorowy będzie pokazywała, w jaki sposób mamy z tym bardzo negatywnym zjawiskiem walczyć.

Tak jak pan poseł mówił, zdefiniowaliśmy tam konkretne kierunki działania. Realizacja tych wszystkich segmentów poszczególnych kierunków warunkuje poprawę sytuacji. Oczywiście możemy się skupić na jednym z tych kierunków, ale bez wielosektorowej, wieloobszarowej działalności wielu różnych instytucji nie osiągniemy tego celu, jakim jest poprawa sytuacji Polaków, którzy doświadczyli choroby nowotworowej. Bardzo ważne są oczywiście kwestie związane z inwestycjami dotyczącymi rozwoju. Tak, to bardzo ważne rzeczy.

Dlatego też jest strategia, która mówi o pewnej hierarchii struktury, jeżeli chodzi o organizację systemu opieki nad pacjentami onkologicznymi. Ma powstać narodowe centrum onkologii oraz regionalne centra onkologii - kolejne podmioty, które będą wykonywały - przy współpracy w pionie i w poziomie - różnego rodzaju świadczenia na rzecz pacjentów onkologicznych.

Te kryteria muszą być ustanowione, muszą być przestrzegane i brane pod uwagę przy wydatkowaniu środków publicznych.

Bez edukacji młodych pokoleń, bez edukacji dorosłych, bez zmiany stylu życia, nawet najnowsze technologie (Dzwonek), najnowsze rozwiązania nie spowodują, że wskaźniki przeżywalności będą lepsze niż w innych krajach europejskich.

Zapraszam pana posła Stanisława Żuka do zadania pytania dodatkowego. Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo!

Kiedy zmienił się dyrektor, zmieniło się podejście. Szanowni Państwo!

Niestety, kontraktu nie było.

Podmiot, który ma zamiar udzielać świadczeń i spełnia, podkreślam, spełnia wszystkie warunki, może być wybrany w trybie konkursu ofert. W Wysokiej Izbie został przegłosowany zapis i Narodowy Fundusz Zdrowia wstrzymał kontraktowanie świadczeń. Dopiero teraz, w październiku, na ostatnim posiedzeniu Sejmu, Sejm znowelizował tę ustawę i w tej chwili odwieszane są postępowania konkursowe. Tam, gdzie jest to niezbędne, fundusz, po przeanalizowaniu potrzeb zdrowotnych, odrębności, jeżeli chodzi o kwestie epidemiologiczne. To jest też uwarunkowane nasyceniem danego rodzaju świadczeniami na danym obszarze.

Takie kryterium nie jest brane pod uwagę.

Przeanalizujemy. Dziękuję bardzo, pani minister. Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie skierowane do ministra klimatu i środowiska w sprawie programu „Czyste powietrze” 2.0 przygotowane jest przez posłów Barbarę Bartuś, Waldemara Andzela oraz Jacka Osucha z Prawa i Sprawiedliwości. Jako pierwsza pytanie zada pani poseł Barbara Bartuś. Dziękuję. Panie Ministrze!

To program skierowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy. Założenia tego programu w moim przekonaniu były znane, są znane, bo w 2018 r. przeprowadzone były liczne spotkania, swego rodzaju szkolenia. Program „Czyste powietrze” przewiduje dofinansowanie m.in. na wymianę stałych źródeł ciepła, tj. pieców, kotłów na paliwa stale, docieplanie budynków, przegród budynków, wymianę okien i drzwi, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalację odnawialnych źródeł energii i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dofinansowanie może zostać wypłacone bezpośrednio wykonawcy. Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tys. zł. Maksymalnie można uzyskać 90% z 53 tys. zł, czyli blisko 48 tys. zł w ramach jednego dofinansowania. Pozostałe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia przekraczające kwotę dotacji mogą być dofinansowane w formie pożyczki, ale też tylko do wysokości 53 tys. zł. Wysokość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Biorąc to wszystko pod uwagę, pragnę zapytać pana ministra, jak wygląda obecnie stan wdrożenia programu, na czym dokładnie polega druga odsłona programu „Czyste powietrze” i co zostało zmienione w kontekście wysokości poziomu dofinansowania dla najuboższych. Dziękuję bardzo, pani poseł. Odpowiedzi na postawione pytanie udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu pan minister Ireneusz Zyska. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Poseł! Bardzo dziękuję za pytanie dotyczące programu „Czyste powietrze” Muszę powiedzieć, że ten priorytetowy program rządu, który jest związany z walką o czyste powietrze czy też zabieganiem o lepszą jakość życia polskich obywateli zarówno w miastach, jak i na całym terytorium kraju, z termomodernizacją, wymianą źródeł ogrzewania, wymianą stolarki okiennej, z możliwością montażu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, stwarza ogromne możliwości w zakresie podniesienia poziomu jakości życia mieszkańców.

Stąd też podjęliśmy działania związane, po pierwsze, z rozszerzeniem programu na osoby najuboższe, na osoby, które osiągają dochód miesięczny netto do 1400 zł na głowę w gospodarstwie domowym albo do 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym. Chodzi o to, aby takie osoby, które dysponują niestety mniejszymi dochodami, mogły również skorzystać z programu „Czyste powietrze”, uzyskując większe wsparcie.

W porównaniu do innych czynności wykonywanych przez gminę w ramach programów rządowych jest to wysoka rekompensata za tę jednorazową czynność. Osoby takie mogą uzyskać dofinansowanie aż do 37 tys. zł, co stanowi według różnych przeliczników dotację w wysokości do 60% poniesionych kosztów na termomodernizację, na wymianę źródła ogrzewania. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu rozwiązaniu, które weszło w życie 21 października br. zdecydowanie większa liczba mieszkańców, którzy do tej pory nie mogli sięgnąć po środki z programu „Czyste powietrze”, będzie mogła je wykorzystać dla poprawy standardu efektywności energetycznej swojego miejsca zamieszkania. Trzeba również powiedzieć, szanowni państwo, że doskonałe narzędzie wprowadził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postaci strony internetowej, która dysponuje takim formularzem zgłaszania wniosku przez Internet. Ten wniosek jest skojarzony także z programem „Mój prąd” Możemy za pomocą jednego formularza aplikować o środki zarówno z programu „Czyste powietrze”, jak i z programu „Mój prąd” Dzięki temu każdy zainteresowany może samodzielnie wyliczyć, jakiej wartości dotację otrzyma. Również ważna informacja jest taka, że od 2019 r. nie płacimy podatku z tytułu uzyskania dotacji z programu „Czyste powietrze” Również ważna informacja: beneficjenci mogą odliczyć od podstawy opodatkowania tzw. ulgę termomodernizacyjną do wysokości 53 tys. zł.

Szanowni Państwo! Szanowna Pani Poseł! Program „Czyste powietrze” jest emanacją i skutecznym wymiarem działań rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, który jakość powietrza w Polsce przyjął jako priorytet.

To ustawa, którą zmienia się trochę program „Czyste powietrze”, modyfikuje się program „Stop smog”, tworzy się Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. Dzięki temu uzyskujemy nowe narzędzia. Może jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć, bo te rozwiązania wejdą w życie w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy po podpisie pana prezydenta, ale to jest również bardzo ważne do tego, abyśmy rozszerzyli oddziaływanie środków, które zostały przeznaczone na program „Czyste powietrze” Dziękuję bardzo, panie ministrze. Będzie pan jeszcze miał okazję o tym powiedzieć, bo dostanie pan 3 minuty po pytaniu dodatkowym. Chciałem państwa serdecznie przywitać. W tym czasie, chciałem obiecać, nie będę wzywał Straży Marszałkowskiej, nie będę arogancki, [[Oklaski]] nie będę nikogo obrażał. Nikogo nie będę też wykluczał.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Program „Czyste powietrze” jest niezwykle ważny dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, dla partii Prawo i Sprawiedliwość, ale w szczególności - dla wszystkich obywateli Polski, którzy od dawna na niego oczekiwali, bo to jest największy program ekologiczny. Mam pytania. Czy przewiduje się stworzenie programu „Czyste powietrze” dla budynków wielorodzinnych: bloków, kamienic itp. Jakie są dalsze plany rozwoju tego programu? Czy nie ma żadnych zakłóceń w realizacji tego niezwykle ważnego programu?

Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Panie ministrze, zapraszam. Wysoka Izbo!

Po pierwsze, został utworzony Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji, który jeszcze bardziej rozszerza możliwość skorzystania ze środków z programu „Czyste powietrze” przez osoby gorzej sytuowane finansowo, które co prawda mają zdolność kredytową, ale nie posiadają żadnego majątku, żadnego zabezpieczenia, żeby wziąć kredyt bądź pożyczkę w banku. W ramach tego rozwiązania zgłaszają się banki komercyjne, które formułują własne programy na preferencyjnych warunkach, o zdecydowanie obniżonym oprocentowaniu, które dedykują właśnie takim osobom. Ten utworzony Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji, którego dysponentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, spowoduje, że banki komercyjne będą mogły udzielać tych pożyczek na preferencyjnych warunkach. Czyli rozszerzamy katalog możliwości skorzystania ze środków finansowych dla osób, które chcą dokonać poprawy standardu swojego miejsca zamieszkania. Drugi element. Tutaj odpowiem na pytanie pana posła Waldemara Andzela w kontekście pytania o budynki wielorodzinne.

To oczywiście nie wszystko, gdyż w tej chwili przygotowujemy program pilotażowy na razie, ale dedykowany dla gmin o największym zanieczyszczeniu powietrza. Taką gminą, w której byliśmy niedawno, w sierpniu chyba, pod koniec sierpnia, z panem ministrem klimatu i środowiska, panem Michałem Kurtyką, jest Pszczyna. Tam zostanie w przyszłym roku, 2021 r., uruchomiony (Dzwonek) program pilotażowy, który będzie dedykowany dla wszystkich gmin o największym zanieczyszczeniu powietrza - program mający w swoim zamierzeniu w ciągu 2, maksymalnie 3 lat eliminację zanieczyszczeń powietrza poprzez w 100% wymianę źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne. Ponadto trzeba powiedzieć, że bardzo ważny element we wczoraj przegłosowanej przez Wysoką Izbę ustawie to utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. To narzędzie, które pozwoli zinwentaryzować w skali całego kraju potrzeby termomodernizacyjne i środki z programu „Czyste powietrze” czy też innych programów, takich jak „Stop smog”, częściowo w skojarzeniu, ponieważ mamy możliwość wspólnego aplikowania, jeśli chodzi o program „Mój prąd”, skierować tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne, abyśmy tych środków nie marnowali, bo są to środki publiczne, powinny być jak najlepiej wykorzystane, najbardziej efektywnie. Szanowni państwo, jestem przekonany, że te rozwiązania, które już funkcjonują i które wejdą w perspektywie. Jakby pan mógł powolutku, ale nie spiesząc się za bardzo, zmierzać ku końcowi, to byśmy byli bardzo zadowoleni. Kończąc, chciałem właśnie powiedzieć, że już te rozwiązania, które w tej chwili funkcjonują w ramach drugiej odsłony programu „Czyste powietrze”, która została wdrożona w dniu 21 października, jak również te, które Wysoka Izba przyjęła w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która to ustawa wejdzie za mniej więcej 30 do 40 dni, 30 dni od opublikowania po uzyskaniu pod aktem prawnym podpisu pana prezydenta, jak też te, o których mówiłem, w ramach działań skierowanych do miast o największym zanieczyszczeniu powietrza, głównie na Górnym Śląsku, i tutaj pierwszym miastem, to jest już ustalone, jako miasto pilotażowe będzie Pszczyna - dają wielką nadzieję na skokowy postęp w zakresie uzyskania poprawy jakości powietrza w Polsce. Jestem przekonany, że te narzędzia pozwolą w większym stopniu wykorzystać tę wielką pulę środków, którą rząd Polski przeznaczył na walkę ze smogiem, a przypomnę, jest to w horyzoncie 11 lat kwota 103 mld zł. Dziękuję uprzejmie, panie ministrze. Chciałem panu powiedzieć, że przekroczył pan swój czas 3 minuty, ale tak błyskotliwej, tak fantastycznej i tak pełnej treści wypowiedzi dawno nie słyszeliśmy. Dziękuję w imieniu Sejmu polskiego. Proszę państwa, pan poseł Sławomir Nitras i pani posłanka Barbara Nowacka postanowili zadać pytanie w sprawie rządowych planów pomocy branżom: gastronomicznej, rozrywkowej, fitness i weselnej, narażonych na bankructwo w wyniku gwałtownego zamknięcia lub ograniczenia ich działalności w ramach obostrzeń związanych z pandemią, a także planowanego wsparcia dla osób zatrudnionych w tych branżach. Odpowie na to pytanie podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, pani minister Olga Semeniuk, którą serdecznie witamy. Zgodzi się pan, że mówienie o pomocy rządu w kontekście zamykanych branż, m.in. branży gastronomicznej, to duże nadużycie albo grzeczność pana marszałka. 2 tygodnie temu prosiliśmy o to, żeby rząd przedstawił harmonogram działań w związku z pandemią. Wszyscy widzieliśmy, że sytuacja jest bardzo trudna, idzie ku złemu, że nie przygotowaliście nas na jesienną falę pandemii. Prosiliśmy o to, żeby powiedzieć, co będziecie zamykać, czy będziecie zamykać. Premier mówił, że ma wszystko pod kontrolą, zwalczył koronawirusa. I przyszedł zeszły czwartek, kiedy m.in. branża gastronomiczna, branża fitness dowiedziały się, że od soboty ich zamykacie - od soboty. Dowiedzieli się, że za 24 godziny mają zamknąć swoją działalność.

Do grudnia zwolnią 200 tys. pracowników i zamknie się do grudnia 7 tys. barów, restauracji, pubów. Co proponujecie? Zamknęliście ich z dnia na dzień. Dzisiaj media donoszą, że ruszyła Krajowa Administracja Skarbowa, że zaczynacie rozliczać i kontrolować przedsiębiorców, którzy dostali pierwszą pomoc. Teraz tym, których zamknęliście z dnia na dzień, zaproponowaliście ulgę w ZUS-ie na miesiąc - na miesiąc.

Co to jest za pomoc? Ponad 1000... Pan Marczak. Nie pomagacie, kontrolujecie, odbieracie. Nie zamykacie szkół, bo mówicie, że koszty dla gospodarki są ogromne. A co z kosztami dla gospodarki, kiedy w tej branży funkcjonuje 70 tys. firm? Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani minister, zapraszam. Panie Marszałku, również serdecznie witam! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Panie pośle, chciałabym odpowiedzieć, zaczynając od tematu COVID-19 i tego, że działamy w ekstraordynaryjnym tempie, dość szybko informując, kilka dni przed, branże o tym, że będą na jakiś czas w minilockdownie. Chętnie umówimy się z tym wirusem, żeby poczekał 2 tygodnie na to, żebyśmy mogli przygotować procedury zamknięcia branż.

A teraz fakty z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Od marca tego roku doprowadziliśmy do sytuacji, w której bezrobocie plasuje się na poziomie 6,1, jest najniższe w Europie. Chodzi o to, abyście państwo też mieli to na uwadze, dlatego że to nie wy się spotykacie z największą częścią przedsiębiorców, tylko właśnie nasz resort. Panie pośle, proszę mi nie przerywać. 19 października tego roku - spotkanie z branżą handlową. Natomiast chciałabym, żeby pan wysłuchał mojej odpowiedzi do końca, bo czekacie na. Mam do państwa taką prośbę: wysłuchajmy pani minister.

Ze wszystkimi branżami się spotkaliśmy. Przyjęliśmy priorytety ich działań, jak również czynniki, które będą pomagały im i wspierały ich w gospodarce. Przeanalizowaliśmy to międzyresortowo, szczególnie biorąc pod uwagę PFR, ministerstwo finansów i inne podmioty, które są w to zaangażowane. Tarcza branżowa to pakiet wsparcia wypracowany w reakcji na drugą falę pandemii dla branż, które najmocniej odczuły jej skutki. To projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z nowych instrumentów skorzysta, panie pośle, szanowni państwo, 200 tys. firm zatrudniających ponad 372 tys. pracowników. Koszt wsparcia wyniesie prawie 2 mld zł. Środki będą pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. O wsparcie będą mogły ubiegać się branże: gastronomiczna, rozrywkowa, targowa, weselna, fitness, sprzedaż detaliczna, targowiska, bazary. Trudno precyzyjnie dokonać podziału środków pomiędzy branżami. Szereg z tych branż się przenika, np. branża weselna z gastronomiczną czy rozrywkową. Kluczowe środki wsparcia to: zwolnienie ze składek ZUS za listopad - warunkiem jest, aby przychód w listopadzie był niższy o 40% co do roku - świadczenie postojowe za listopad i mikrodotacja w wysokości 5 tys. zł dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Warunkiem jest, aby przychód był niższy o 40%. Chciałabym też podkreślić, że zmniejszyliśmy to kryterium, jeżeli chodzi o procentowy spadek obrotów: z 75%, które były przewidziane w tarczy turystycznej, do 40%. Mikrodotacja dla mikro- i małych przedsiębiorców jest przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacja podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikro- lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Powyższe instrumenty są kierowane do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność oznaczoną kodami PKD, określonymi w ustawie. Przy czym w przypadku postojowego liczba kodów w procedowanej ustawie jest mniejsza, gdyż część z nich pokrywa się z kodami PKD zawartymi w tzw. tarczy turystycznej. O tym mówił wczoraj pan premier Mateusz Morawiecki. Co istotne, projekt przewiduje możliwość przedłużenia tych form wsparcia poprzez stosowne rozporządzenie Rady Ministrów. Decyzje w tym zakresie będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji. Warto też podkreślić, że dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, która uzupełnia tarczę antykryzysową. Pomoc przeznaczona może być wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej w związku z realizowaną restrukturyzacją. Na pomoc firmom w kryzysie jest do dyspozycji 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat. Operatorem tej pomocy jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Panie Pośle! Bardzo często pojawiają się takie zarzuty: dlaczego zamknęliście aquaparki, dlaczego siłownie, dlaczego gastronomię, dlaczego w takim tempie? Wirus się rozwija nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Jeśli chodzi o transmisję wirusową, to są branże, w których skupia się największa liczba osób, w których nie możemy zabezpieczyć noszenia maseczek, w których są skupiska osób. To nie jest tak, że rząd polski chciał od razu zamykać gastronomię, tylko chciał doprowadzić, panie pośle, do sytuacji, w której jednak tym wąskim korytarzem będziemy się przesuwać w minilockdownach, ale nie przy całkowitym zamknięciu gastronomii. Niestety, sytuacja epidemiczna w kraju nam na to nie pozwoliła. Dlatego postanowiliśmy zrobić to na jakiś czas - na razie mamy nadzieję, że to będą 2 tygodnie. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja będzie się zmieniała.

Dziękuję.

że to pani jest członkinią rządu i to od was obywatelki i obywatele wymagają rozwiązań. A kiedy my przynosimy propozycje, państwo macie taki fantastyczny arogancki sposób wyśmiewania, wykpiwania i niesłuchania. Pani urządza sobie drwiny, proponuje, żeby dzwonić do wirusa, a nasze pytanie jest bardzo proste: Jak się przygotowaliście? Były te warianty? Poinformowaliście przedsiębiorców? Zamykacie kluby fitness, a szkoły tańca mogą działać. Zamknęliście restauracje, ale restauracje hotelowe mogą działać. To jest ten regularny plan przygotowania?

I to ma im pani do powiedzenia? To ma pomóc pracownikom? Gdzie w tym wszystkim zgubiliście bardzo ważną rzecz, rynek pracy? Pani sieje tutaj propagandę sukcesu, opowiadając o bezrobociu na poziomie najniższym w Europie, na świecie i o tym, jak cały świat nam zazdrości, a zapomina pani, że bardzo wiele osób w tej branży również dorabiało i że całe bezrobocie też nie chwyta ludzi pracujących dorywczo, nie chwyta tych takich pojedynczych przedsiębiorców. Pani minister, zapraszam.

Jeżeli chce pani uzyskać informację, ile kodów PKD zostało w tym uwzględnionych, to oczywiście to przedłożymy. Przygotowanie protokołów bezpieczeństwa przez ówczesny resort rozwoju, odmrożenia: pierwsze, drugie, trzecie i czwarte, jeżeli chodzi o gospodarkę, przygotowanie tych branż do tego, żeby były odmrożone, jak również szybkie tempo działań w kontekście obecnej tarczy. Nigdy w życiu ani Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, ani polski rząd w żaden sposób nie lekceważyły przedsiębiorców, czego dowodem jest dialog branżowy, czego dowodem są codzienne, cykliczne spotkania z przedstawicielami poszczególnych branż, którzy bardzo chętnie spotykają się z nami. Nie wiem, czy tak samo z panem posłem czy z panią poseł chętnie się spotykają, natomiast z nami spotykają się chętnie. Przedstawiają swoje argumenty, swoje warianty dotyczące chociażby targowisk czy branży handlowej, czy branży hotelarskiej. Pragnę też przypomnieć, że jeżeli chodzi o branżę hotelarską, to właśnie wcielamy w życie przeobrażanie się hoteli w izolatoria, co będzie dodatkowym napędem finansowym. Rząd jest od podejmowania decyzji, rząd jest od przedstawiania różnego rodzaju rozwiązań - pełna zgoda, pani poseł - ale to wy jesteście od tego, aby nie doprowadzać do sytuacji buntów ulicznych, eskalacji konfliktu.

To jest ta solidarność i odpowiedzialność społeczna, o której bardzo często państwu mówimy, i pewnie musimy to definiować jeszcze wiele razy, odpowiedzialność rozłożona pomiędzy pracownika, pracodawcę i rząd. Oczekujemy konkretnych rozwiązań punktowych, branżowych, po to abyśmy mogli ten najgorszy okres przejść. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dowiedzieliśmy się, czego posłowie oczekują od rządu i czego rząd oczekuje od posłów. Pan poseł Piotr Kaleta z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zada pytanie w sprawie stopnia zaawansowania prac przy projektowaniu kolei dużych prędkości i wpływu pandemii na realizację tego projektu. Odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan minister Marcin Horała. Bardzo proszę, panie pośle. A posłom Platformy Obywatelskiej dziękuję serdecznie za obecność. Wysoka Izbo! Docierają do nas informacje, od tego chciałbym zacząć, że oto dzisiaj o godz. 17 na Jasnej Górze - lewicowy potop. Skrajna lewica, która wypycha przed siebie dziewczynki, młode osoby, które nie do końca rozumieją, o co w tym chodzi, chce dokonać bezczelnego ataku na duchową stolicę Polski, na Jasną Górę. Oczywiście nie może być zgody na to, żeby takie działania miały miejsce. Przeżyliśmy potop szwedzki, przeżyjemy i potop lewacki.

Panie pośle, uprzejmie pana informuję, że jest pan wyłączony i pana nie słychać. Więc teraz pan posłucha marszałka Sejmu, który ma taką samą pozycję jak marszałek Terlecki. Niech pan się zajmie zadaniem pytania, bo po to pan tu został wezwany. Jak pan nie ma ochoty tego zrobić, proszę zejść z mównicy. Proszę bardzo. W związku z tym chciałbym, żeby jeszcze raz to wybrzmiało: dzisiaj trzeba stanąć w obronie Jasnej Góry. Jeszcze raz panu mówię, że ma pan 15, 13, 12, 11, 8 sekund. Proszę bardzo. Panie marszałku, to jest bezczelność z pana strony, co pan zrobił, ponieważ nie. Dziękuję serdecznie panu. Dziękuję bardzo.

Wie pan, na czym ona polega? Czy pan się spodziewa, że ktoś z pana obozu politycznego by coś takiego zrobił? Niech pan się uczy. Zapraszam pana.

Wszystko to odczuwa polska gospodarka.

Czy on w dalszym ciągu funkcjonuje?

W jaki sposób w tej chwili te sprawy się układają? Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję serdecznie. Proszę pana, nie sprowokuje mnie pan.

Panowie posłowie, ja sobie dam radę, naprawdę.

Byłbym wdzięczny. Panie ministrze. Czy jest pan minister? Niech pan wchodzi. Proszę bardzo.

Bardzo proszę, panie ministrze. Program inwestycyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego pod względem planowanych nakładów to w 3/4 jest program inwestycji kolejowych. Budowa systemu kolei dużych prędkości, tych tzw. szprych, to jest odwołanie do teorii piasty i szprych jako modelu systemu komunikacyjnego, który dla kraju wielkości i kształtu Polski jest optymalny.

Tak to jest, że w czasach spowolnienia lepiej, szybciej i łatwiej przeprowadza się inwestycje. Wykonawcy częściej szukają zamówień, dają lepsze ceny. To w czasach przegrzania koniunktury, wtedy, kiedy gospodarka jest bardzo rozpędzona, często trudno znaleźć wykonawców, albo oferują oni ceny powyżej kosztorysów. Tą najważniejszą w tym roku było przygotowanie strategicznego studium lokalizacyjnego, czyli formy studium korytarzowego dla całego nowego systemu komunikacyjnego Polski. W toku konsultacji społecznych studium zgłoszono 140 tys. uwag. W przytłaczającej większości nie dotyczyły studium korytarzowego, tylko przykładowych przebiegów linii. Te uwagi będą wykorzystane na etapie, kiedy te przebiegi będą przesądzane. Pierwszy etap, który został skierowany do realizacji, który trwa obecnie, to etap inwentaryzacji środowiskowej będącej najważniejszym elementem przygotowania do uzyskania decyzji środowiskowej.

W kolejnych latach będą uruchamiane kolejne procesy inwestycyjne. To wtedy będą przesądzane konkretne, dokładne przebiegi mieszczące się w szerokich korytarzach transportowych, które zostały zdefiniowane na poziomie konsultacji strategicznego studium lokalizacyjnego.

Wspomnijmy chociażby projekt budowy kolei dużych prędkości Praga - Drezno, czy inne programy tego rodzaju. Jak pokazał raport firmy Kearney, renomowanej międzynarodowej firmy audytorskiej, budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, całego tego systemu komunikacyjnego, to 95 tys. nowych miejsc pracy, z czego 80% w sektorze budowlanym.

To 238 tys. miejsc pracy w samym porcie i jego otoczeniu, 290 tys. miejsc pracy w gospodarce, 780 mld wartości dodanej brutto i prawie 1 bln zł wzrostu produkcji w perspektywie do roku 2040.

Polska dzięki programowi inwestycyjnemu CPK może trafić do pierwszej ligi zarówno w wymiarze światowym - pojawi się duże hubowe lotnisko będące ważnym punktem komunikacyjnym na mapie świata - jak i (Dzwonek) w wymiarze krajowym, przez polepszenie dostępności właśnie w systemie szprych, szprych i piasty przez CPK czy przez węzeł kolejowy CPK będą również podróżowali Polacy, którzy będą chcieli przemieszczać się z jednej części kraju do drugiej, niekoniecznie korzystać z lotniska. Powiem, że największym beneficjentem tego systemu wydają się być miasta średniej wielkości, te, które do tej pory są praktycznie wykluczone komunikacyjnie, w ogóle nie mają połączeń kolejowych albo mają bardzo rzadkie i bardzo niewygodne połączenia.

Bardzo dziękuję. Czy pan poseł ma pytanie dodatkowe? Bardzo proszę, panie pośle. Chciałbym się jeszcze dopytać pana ministra, jak wygląda kwestia, jeśli chodzi o koleje wielkich prędkości, stricte dotycząca przebiegu tzw. dawnego igreka. Może dzisiaj igrek to jest, żeby to sprecyzować, kwestia dotycząca rozwidlenia w okolicach Sieradza, które miało iść również w kierunku Kalisza. Jeżeli byłby to kłopot, to oczywiście prosiłbym pana ministra o jakąś odpowiedź na piśmie. Pana marszałka chciałbym jeszcze pouczyć, że dobrze by było, żeby marszałek nie miał na twarzy pewnych emblematów, które mogą sugerować podniesienie wysokiego napięcia. Może pan o tym nie wiedzieć, ale nie dziwię się. Poprosimy pana ministra Horałę. Panie pośle, chciałem panu powiedzieć, że chciałem pana bardzo, bardzo uprzejmie przeprosić, jeżeli cokolwiek w moim zachowaniu wpłynęło na to, że pan poczuł dyskomfort. Jest mi z tego powodu bardzo przykro.

Dziękuję bardzo. Dziękuję. Najpierw tytułem uzupełnienia jeszcze jednego etapu inwestycji, o którym nie wspomniałem. Oczywiście toczy się również proces uzyskiwania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko całego programu inwestycyjnego. On będzie zakończony najdalej w styczniu przyszłego roku, co pozwoli, da możliwość ubiegania się o środki europejskie dla wszystkich projektów z tego programu. Jestem przekonany, że będzie to taką jaskółką, która czyni wiosnę, i w następnych perspektywach spore środki europejskie na ten program będziemy pozyskiwać. Dziś na posiedzeniu Rady Ministrów staje uchwała o wieloletnim programie finansowym Centralnego Portu Komunikacyjnego, która zapewni w perspektywie do roku 2023, czyli na prace projektowe, przygotowawcze, wykup gruntów i rozpoczęcie inwestycji, kwotę ponad 13 mld zł, co niezwykle istotne, nie obciążając tym budżetu państwa, nie będzie żadnych kosztów, ani złotówki, dla budżetu państwa. Program Centralnego Portu Komunikacyjnego to jest również w pewnym aspekcie wielki program pozyskiwania do Polski kapitału z zewnątrz, środków europejskich, środków komercyjnych na dobre inwestycje, wpisujące się w politykę europejską, jak również po prostu komercyjnie opłacalne, tak jak duże lotnisko hubowe.

Później ten naturalny etap uzyskiwania decyzji środowiskowej będzie również etapem konsultacji społecznych, takich pogłębionych, na miejscu, w gminach, i ustalania ostatecznego przebiegu. Tak to jest, że do momentu uzyskania decyzji środowiskowej trzeba pokazywać przynajmniej trzy warianty. To decyzja środowiskowa przesądza, jaka jest ostateczna lokalizacja. Panie ministrze, dziękuję bardzo, bardzo serdecznie.

W imieniu Ministerstwa Finansów będzie odpowiadała pani minister Anna Chałupa. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Minister! Od października zaczyna obowiązywać nowy plik JPK_VAT z deklaracją. Jeden plik ma zastąpić dotychczas składane oddzielnie deklaracje. Jednak częste zmiany powodują to, że przedsiębiorcy czują się niepewnie, szukają informacji o nowych rozwiązaniach. Do tego dochodzą kontrole z urzędu skarbowego, które mają negatywny wpływ na płynność działania firmy. Dotyczy to szczególnie tych najmniejszych firm: mikro-, małych firm, które same się rozliczają.

Proszę o taką informację, chodzi o informacje, które są chociażby na stronie ministerstwa, czy ten nowy system ewentualnie będzie generował po stronie przedsiębiorców korzyści.

Dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Zapraszam panią minister. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który składa się z dwóch części: ewidencji VAT i deklaracji VAT.

Nowy plik będzie obejmował zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT, pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 czy VAT-7K oraz dodatkowe dane. JPK_VAT z deklaracją będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej, więc to jest już pierwsze uproszczenie, a także będzie go można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi. Po złożeniu JPK_VAT z deklaracją podatnik będzie mógł pobrać urzędowe poświadczenie odbioru danych. Ministerstwo Finansów udostępni przedsiębiorcom bezpłatne narzędzia, które pomogą im przygotować, podpisać i wysłać pliki JPK_VAT z deklaracją. Udostępnione zostaną: formularz interaktywny, tzw. bramka, i nowa wersja aplikacji e-mikrofirma. Formularz interaktywny będzie prostym w obsłudze narzędziem webowym, które wymaga połączenia z Internetem. Zastąpi dotychczasowy plik w formacie CSV, który był dość niewygodny, a z formularza będą mogli korzystać także podatnicy posiadający kontrahentów zagranicznych, co jest nowością. Jeśli chodzi o nową aplikację e-mikrofirma, to umożliwi ona wystawianie i zapisywanie faktur krajowych, stworzenie ewidencji VAT oraz wygenerowanie i wysyłanie plików JPK_VAT. Nowa wersja aplikacji zastąpi jej dotychczasową wersję desktopową. Do aplikacji będzie się można zalogować za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Dotychczasowi użytkownicy tego narzędzia będą mogli płynnie przejść na użytkowanie nowszej wersji z rozbudowanymi funkcjonalnościami dzięki wbudowanej opcji importu, eksportu danych. Więc nowe narzędzie będzie obsługiwać także historyczne dane. Jeśli chodzi o kanały komunikacji, to elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie ministra finansów, inwestycji i rozwoju z dnia 15 października 2019 r. oraz opracowany na jego podstawie wzór schemy JPK_VAT, który jest opublikowany w centralnym rejestrze wzorów dokumentów elektronicznych na ePUAP. Ministerstwo Finansów na stronach portalu podatkowego na bieżąco informowało o pracach nad wprowadzeniem nowego rozwiązania. Wszelkie informacje są cały czas dostępne na portalu podatkowym. Ostatnie komunikaty przypominające o nowym pliku zamieszczono na stronach Ministerstwa Finansów na dzień przed wprowadzeniem tego rozwiązania, jeszcze 30 września 2020 r. Informacje o nowym rozwiązaniu z odesłaniem do portalu podatkowego Ministerstwo Finansów od IV kwartału 2019 r. zamieszcza także w kierowanych do przedsiębiorców z poziomu centralnego powiadomieniach e-mail lub SMS-ach, w momencie kiedy identyfikujemy jakieś niezgodności w dotychczasowych rozliczeniach VAT. Jednocześnie, oczywiście dzięki współpracy z mediami, informacje o nowym JPK_VAT od końca 2019 r. systematycznie pojawiają się w różnego rodzaju artykułach prasowych. Jeśli chodzi o korzyści, to najważniejszą korzyścią jest to, że przedsiębiorca, zamiast - tak jak jest obecnie - składania odrębnie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz z załącznikami i odrębnie informacji JPK_VAT będzie przesyłał jeden plik JPK_VAT, realizując łącznie dwa obowiązki. Nie będzie potrzeby generowania dwóch plików, składania dwóch podpisów, dokonywania dwóch wysyłek i dwukrotnego oczekiwania na tzw. UPO. Zostanie także dzięki temu ograniczona liczba kontroli podatkowych i postępowań oraz skróci się czas wykonywania czynności kontrolnych. Każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika. Zapewni nam to właśnie ten system. Dodatkowo urząd skarbowy będzie szybciej mógł weryfikować zwroty VAT z uwagi na równoczesne przesyłanie przez podatników deklaracji i szczegółowych informacji z ewidencji. Dziękuję. Ja również pani bardzo serdecznie dziękuję. O pytanie dodatkowe proszę pana posła Kazimierza Smolińskiego z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dosyć szczegółowo pani minister przedstawiła informacje związane ze zmianami.

Myślę, że kwestia, że to jest uproszczenie dla przedsiębiorców, to nie ulega wątpliwości. Natomiast jakby pani minister mogła jeszcze raz też korzyści, które wynikają z tego po stronie Skarbu Państwa. Czy to jest element uszczelniania systemu podatkowego? Jednolity plik kontrolny właśnie w tej podwójnej wersji, który do tej pory obowiązywał, teraz jako jednolity - czy można też powiedzieć, że on jest jakimś elementem do wprowadzania w przyszłości centralnej ewidencji faktur, bo myślę, że do tego powinniśmy zmierzać. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Pani minister, zapraszam. Panie Marszałku! Panie Pośle! Oczywiście korzyści z elektronizacji sposobu składania deklaracji są jak najbardziej dla nas ogromnym plusem, gdyż dzięki nim będziemy mogli wykluczać wszelkie ryzyka uwikłania w oszustwo podatkowe.

Oni dzięki temu będą mogli lepiej zarządzać swoimi przedsiębiorstwami. Także sam fakt, że ograniczymy liczbę kontroli podatkowych i postępowań, czyli skrócimy także czas wykonywania czynności sprawdzających oraz kontrolnych, to też jest oddech dla przedsiębiorców. Dzięki temu nie będziemy musieli fizycznie do nich przychodzić, będziemy mogli ich obsługiwać zdalnie.

Oczywiście będziemy myśleć o dalszych usprawnieniach, łącznie z rejestrem faktur centralnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Teraz poproszę pana posła z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Mariusza Trepkę o zadanie pytania w sprawie planu wprowadzenia nauki zdalnej w całym kraju. Odpowiadała będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pani minister Marzena Machałek. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo! Jak wiemy, od poniedziałku naukę zdalną mamy we wszystkich zakresach szkół, od szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I-III, po szkoły średnie i uczelnie wyższe. Moje pytanie jest bardzo konkretne: Jakie rozwiązania rząd przygotował do nauki zdalnej w zakresie szkół specjalnych, zawodowych i placówek z kształceniem ustawicznym?

Oczywiście warto powiedzieć, że kształceniem ani hybrydowym, ani zdalnym nie chcieliśmy objąć dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczących się w szkołach specjalnych, w specjalnych ośrodkach edukacyjnych, a także wychowanków MOW-ów i MOS-ów, dlatego też pozostawiliśmy dowolność, czyli pozostawiliśmy to do decyzji dyrektora, który ocenia bezpieczeństwo szkoły pod względem kadrowym. Nauka w szkołach specjalnych się odbywa i to jest bardzo ważne, bo 33 tys. dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczy się w 982 szkołach specjalnych. Chcę powiedzieć, że też zadbaliśmy o to, żeby odbywały się zajęcia rehabilitacyjno-wychowawcze, rewalidacyjno-wychowawcze, a także o to, co dla nas jest ważne - żeby nie zaprzestać wczesnego wspomagania dzieci zagrożonych niepełnosprawnością bądź dzieci z niepełnosprawnościami. Natomiast oczywiście tutaj zostawiamy do decyzji rodziców i decyzji dyrektorów szkół, placówek, aby takie zajęcia, których brak może skutkować przez całe życie dzieci, były podejmowane z rozwagą, z rozsądkiem, po ocenie zagrożenia. Natomiast jeśli chodzi o szkoły branżowe i zawodowe, to mam bardzo dobrą wiadomość dla państwa, bo po naszej reformie kształcenia branżowego i zawodowego mamy zdecydowaną, bardzo istotną zmianę trendu i mamy już 56,5% absolwentów szkół podstawowych, którzy trafiają do techników i szkół branżowych, i widzimy zdecydowany wzrost naboru do szkół branżowych.

Natomiast chcę powiedzieć, że po okresie wiosennego lockdownu pierwsze decyzje o powrocie do zajęć stacjonarnych dotyczyły przede wszystkim kształcenia praktycznego. Odmrażaliśmy wszystkie zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe, w pierwszej kolejności na kursach zawodowych oraz w ostatnich klasach i semestrach szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Podjęliśmy decyzję, że nie dotyczy to zajęć praktycznych, praktycznej nauki zawodu.

Na pierwszej linii wprowadzania z powrotem dzieci i młodzieży do nauczania stacjonarnego to będą szkoły zawodowe, a szczególnie ostatnie klasy przed egzaminami oraz oczywiście klasy VIII i klasy maturalne. Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy ograniczyć podstawy programowej w kształceniu zawodowym, bo nie można, mając konkretny zawód, zdany egzamin, czegoś w tym zawodzie nie umieć, co odpowiada za bezpieczeństwo, za jakość wykonanej pracy.

Dziękuję. Pani Minister! Jaką pomoc rząd przewiduje dla szkół w zakresie nauki zdalnej? Czy szkoły otrzymają dodatkowy sprzęt w postaci komputerów i tabletów? Jakie środki rząd przeznaczy na tę pomoc? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo często w przestrzeni publicznej są zafałszowane bądź nieprawdziwe informacje.

Mieliśmy dwie transze.

Później była kolejna transza, też prawie 370 mln. To, na co zwróciliśmy uwagę, to 130 mln dla dzieci w pieczy zastępczej. Oczywiście w tej chwili do szkół trafiają komplety i zestawy tabletów, prawie 40 tys. tych zestawów. Do końca roku rozdamy szkołom kolejne 35 mln na zakup komputerów i sprzętu multimedialnego. Już wiemy, i to też premier zapowiedział, że będzie kolejne 300 mln na zakup sprzętu dla szkół.

To bywa czasem niezbędne, czego dzisiaj też doświadczamy w Sejmie, ale w szkole naprawdę bardzo ważny jest kontakt, bardzo ważna jest socjalizacja, ważne jest wspieranie dzieci przez nauczycieli.

Przygotowaliśmy wraz z sanepidem i ministrem zdrowia odpowiednie wytyczne, odpowiednie warianty, które pozwalają na przechodzenie na różne modele w zależności od zagrożenia.

Daliśmy bardzo dużo elastycznych narzędzi dyrektorom przy wsparciu nauczycieli, jeżeli chodzi o programy kształcenia nauczycieli w zakresie umiejętności cyfrowych. Cały czas oczywiście analizujemy wszystkie uwagi, analizujemy wszystkie wątpliwości. Staramy się na bieżąco odpowiadać. Przez system informacji oświatowej dociera to do dyrektorów szkół.

Tak że jesteśmy w każdej chwili do państwa dyspozycji. Dziękuję serdecznie. Następne pytanie zada pani poseł z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Joanna Borowiak, a będzie ono dotyczyło skali realizacji uprawnień do uzyskania dodatku solidarnościowego. Na to pytanie odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pan minister Stanisław Szwed. Wysoki Sejmie! W ramach walki ze skutkami gospodarczymi koronawirusa rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował i wdrożył mechanizmy wsparcia na łączną kwotę ponad 150 mld zł. Wspieramy przedsiębiorców, pracodawców i pracowników we wszystkich obszarach. W czerwcu zostały przyjęte i wdrożone również przepisy adresowane do osób, które w następstwie COVID-19 straciły pracę. Te przepisy dotyczą wszystkich pracowników, z którymi pracodawca rozwiązał umowę o pracę lub jej nie przedłużył i uległa ona rozwiązaniu. Także w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał pierwszych wypłat dla osób, które złożyły wnioski, a te wnioski można było składać do końca sierpnia. Panie Ministrze! W imieniu własnym oraz moich koleżanek, pani poseł Lidii Burzyńskiej i pani poseł Joanny Milczanowskiej, chciałabym pana ministra poprosić o odpowiedź na pytanie: Jaka była skala udzielonego dotychczas wsparcia dla pracowników, którzy w następstwie epidemii koronawirusa stracili pracę? Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, pani poseł. Zapraszam pana ministra. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję pani poseł za to pytanie dotyczące w ogóle funkcjonowania tarczy antykryzysowej, ale tutaj w odniesieniu do tego konkretnego przykładu, jakim jest dodatek solidarnościowy przyznawany w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, warto przypomnieć, że to była inicjatywa pana prezydenta Andrzeja Dudy, który zgłosił ten projekt do Sejmu, a główny cel tego był związany z sytuacją, która była w kwietniu, maju, czyli sytuacją dotyczącą rynku pracy. Niektórzy eksperci wieszczyli, że będzie bardzo wysokie bezrobocie. Do dzisiaj mamy ustabilizowaną sytuację na rynku pracy, ale wtedy też pojawiła się propozycja ze strony pana prezydenta, aby objąć dodatkowym wsparciem te osoby, które z jakichś względów traciły pracę, czyli osoby, które po 15 marca - w momencie gdy zaczęliśmy zwalczać COVID-19 - straciły pracę, aby mogły skorzystać z dodatku solidarnościowego. To było jedno rozwiązanie.

Jeśli chodzi o te rozwiązania, które po raz pierwszy zaproponowaliśmy, bo dodatek solidarnościowy zaczął wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych, było istotne, że w tym rozwiązaniu po raz pierwszy wprowadziliśmy składanie wniosków tylko w systemie elektronicznym.

Wprowadziliśmy system elektroniczny przez PUE ZUS-u, czyli mieliśmy tę możliwość, żeby od razu te środki były wypłacane. ZUS też bardzo mocno zaangażował się w to, żeby pomagać, zakładać profile zaufane.

Istotne jest też to, że dodatek solidarnościowy wlicza się nam do stażu emerytalnego i składka na ubezpieczenie społeczne jest odprowadzana, czyli tutaj też Zakład Ubezpieczeń Społecznych tego dokonuje, a pracownik - w tym przypadku ten, który jest na dodatku solidarnościowym, tak jak w przypadku tego, który jest na zasiłku dla bezrobotnych - na tym nie traci.

Przypomnę, że dodatek solidarnościowy był na miesiące: czerwiec, lipiec i sierpień.

To jest ten podstawowy zasiłek i on w tej chwili wynosi 1200 zł, czyli z tej kwoty 880 zł zasiłek dla bezrobotnych też wzrósł do 1200 zł.

Czyli nie mamy wzrostu bezrobocia.

Cieszę się, że w ten sposób mogliśmy pomóc pracownikom, którzy tracili pracę i przez dodatek solidarnościowy mieli środki na funkcjonowanie. Dziękuję serdecznie, panie ministrze.

Ale to wie pan, to tak idzie po prostu. Pani poseł, bardzo proszę. Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, za ukazanie całego spektrum pomocy rządu Prawa i Sprawiedliwości dla osób, które straciły pracę na skutek epidemii COVID-19, dla osób bezrobotnych. Mam do pana ministra jeszcze prośbę o wskazanie, jakiego rzędu wsparcie zostało udzielone w kraju, z podziałem na województwa i ze szczególnym uwzględnieniem województw: kujawsko-pomorskiego, śląskiego oraz łódzkiego. Nas bardzo interesuje to, jakiej wysokości środki finansowe zostały przekazane dla naszych obywateli jako wsparcie w sytuacji koronawirusa, tak by mogli poradzić sobie finansowo. Dziękuję bardzo. Proszę, panie ministrze. Wysoka Izbo! Pani poseł, jeśli chodzi o to pytanie dotyczące rozbicia dodatku solidarnościowego i wypłat w rozbiciu na poszczególne województwa, to tak jak już powiedziałem, ogólna kwota to było 234 tys. wypłaconych świadczeń na kwotę pond 313 mln zł.

Jeśli chodzi o województwo mazowieckie - ponad 32 tys. wypłaconych świadczeń na kwotę ponad 43 mln zł. Mamy też rozbicie na poszczególne oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowe dane, jeżeli pani poseł sobie życzy, też prześlemy. Dziękuję panu ministrowi. Prawda, że było miło? Super. Marszałek jest inteligentny, to ma kąśliwe uwagi. Proszę państwa, pani posłanka Urszula Zielińska oraz pan poseł Marcin Kierwiński z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska zadadzą pytanie w sprawie przekraczania uprawnień oraz agresywnych działań ze strony Policji w czasie protestów kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To pytanie jest skierowane do ministra spraw wewnętrznych, reprezentuje go sekretarz stanu pan minister Maciej Wąsik, którego witamy serdecznie. Proszę bardzo, pani posłanko. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! To nasz błąd. Panie Ministrze! Z protestującymi na ulicach Warszawy od tygodnia kobietami jestem codziennie i z bliska obserwuję działania policji. Przyznam, że coraz częściej udaje mi się z policją współpracować, deeskalować konflikty i rozładowywać napięte sytuacje. Policja, która pracuje w niezwykle trudnych warunkach epidemii, coraz częściej pokazuje, że jest z obywatelkami i obywatelami, szuka dialogu, robi wiele, żeby łagodzić konfliktowe sytuacje. I za to chciałabym policjantkom i policjantom oraz dowodzącym na ulicach Warszawy i w całej Polsce podziękować. Jednocześnie zaobserwowałam wiele sytuacji, które wskazują na systemowy problem. Policja bywa wykorzystywana jako firma ochroniarska przez skrajnych nacjonalistów. Oto jeden tylko przykład, chociaż mam ich więcej. Niedziela, Krakowskie Przedmieście, przed kościołem św. Krzyża, osiłek z tzw. straży narodowej poleca policjantom, aby wynieśli z podestu przed kościołem starszą kobietę. Na nagraniu słychać, że dowodzący się wzbrania, ale w końcu się poddaje i mówi: My możemy asystować, ale panowie sami znoszą. Na te słowa kilku osiłków ze wsparciem policji popycha starszą panią ze schodów i wyrzuca poza chroniący schody kordon policji. Te przykłady, wszystkie przykłady, które mam z ostatnich dni, opiszę panu ministrowi dokładnie w interpelacji. Ale mam pytanie, panie ministrze: Czy w MSWiA jest przyzwolenie na współpracę z narodowcami, ze skrajną prawicą? Czy zgadza się pan, żeby polska policja była wykorzystywana w taki sposób przez skrajnych nacjonalistów i w taki sposób traciła wiarygodność i zaufanie, które z trudem budowała przez ostatnie 30 lat? Zapraszam pana ministra.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rzeczywiście reprezentuję pana ministra Mariusza Kamińskiego, który jest w kwarantannie. Da Bóg, jutro wynik testu będzie ujemny i będzie mógł powrócić z pracy zdalnej do kierowania bezpośrednio resortem. Chciałem państwa zapewnić, że Mariusz Kamiński kieruje resortem zdalnie, przy pomocy swoich zastępców, jest w stałym kontakcie ze wszystkimi szefami służb podległych MSWiA. Szanowni państwo, w ostatnich dniach przez Polskę przetoczyły się protesty uliczne, którym towarzyszyły niestety oburzające ataki na kościoły, na miejsca kultu. W ostatnich dniach zanotowaliśmy 22 wtargnięcia na msze święte i zakłócenia tychże mszy. Zanotowaliśmy 79 zdewastowanych napisami przez pseudoprotestujących. Zanotowaliśmy 79 zdewastowanych elewacji, często zabytkowych, najczęściej zabytkowych kościelnych budynków, związanych z kultem, ale nie tylko, bo np. zdewastowane zostało ogrodzenie jadłodajni, którą prowadzą siostry zakonne, i obok jest przedszkole, gdzie pojawiły się wulgarne napisy. Dochodziło także, choćby ostatniej nocy, do ataków na policjantów czy też ludzi, którzy stali przy kościołach, żeby pilnować tychże kościołów. To barbarzyństwo, szanowni państwo. Chciałbym powiedzieć, że w związku z tymi wydarzeniami zatrzymano 76 osób w celu postawienia zarzutów karnych. Policja prowadzi ponad 100 postępowań, żeby ustalić innych sprawców tychże zdarzeń - tych, którzy obrażali uczucia religijne, dewastowali lub atakowali policję bądź też inne osoby postronne, a także tych, którzy niszczyli mienie albo np. skakali po prywatnych samochodach zaparkowanych w mieście. Nie ma na to przyzwolenia. Policja reagowała, reaguje i reagować będzie, adekwatnie do sytuacji, na wszelkie akty agresji, na wszelkie ataki na ludzi, na ataki wobec kościołów, na zakłócanie obrzędów religijnych.

W tym kontekście, pani poseł, uważam, że reakcje Policji, które także pani opisywała, były adekwatne do sytuacji i Policja działa w sposób adekwatny i prawidłowy. Nie widzę powodów, dla których mielibyśmy karać policjantów. Trzeba ich nagradzać. Zapraszam pana posła Marcina Kierwińskiego, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Usłyszeliśmy rzecz skandaliczną. Pani poseł pytała o to, jak to się dzieje, że narodowcy zachowujący się w sposób skandaliczny pobili kobietę na Krakowskim Przedmieściu, a pan minister mówi, że to adekwatna reakcja Policji. Rozumiem, panie ministrze, że dla pana adekwatne jest to, że jak biją kobietę, to Policja stoi i nie reaguje. Rozumiem, że to jest dla pana adekwatne zachowanie Policji.

Pan nie został tutaj zaproszony po to, aby opowiadać o tym, jak to dzielnie bronicie kościołów. Pan został tu zaproszony po to, aby powiedzieć, czy będzie pan wyciągał konsekwencje wobec tych policjantów, którzy przekraczają uprawnienia. Na to pan nie potrafi odpowiedzieć. Czyli wszelkie przejawy agresji [[Dzwonek]] pan usprawiedliwia, nie zamierza pan wszcząć postępowań kontrolnych, nie zamierza pan sprawdzić tych sytuacji. To jest skandal. Jeżeli ktoś był skazany przez polski sąd, to chyba nie potrafi rzeczywiście wyciągnąć z tego żadnych wniosków, a pan niestety tak działa. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Panie ministrze, bardzo proszę. Pan poseł Kierwiński po prostu mnie nie zrozumiał. Mówiłem bardzo wyraźnie, że wszelkie ataki agresji będą ścigane przez Policję. Wszelkie akty dewastacji będą ścigane przez Policję. Nieważne, czy to zrobili czarni, żółci, czerwoni, czy biali.

Dziękuję serdecznie za tę wypowiedź. Proszę państwa, zamykamy ten punkt. Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie dostępności lekarzy ginekologów, gabinetów ginekologicznych, w tym dla kobiet z niepełnosprawnościami, badań prenatalnych i zabiegów przerywania ciąży, o której przedstawienie wnosił Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia) Przypominam również, że przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 5 minut. Wystąpienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty. Na zakończenie dyskusji głos zabierają kolejno przedstawiciel wnioskodawców oraz przedstawiciel Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 5 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia przedstawiciela Rady Ministrów. Czas przeznaczony na rozpatrzenie punktu: Informacja bieżąca nie może być dłuższy niż 90 minut. Bardzo uprzejmie proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców panią posłankę Marcelinę Zawiszę. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Wiceminister! Po skandalicznym wyroku Trybunału Konstytucyjnego wnoszę o informację bieżącą od ministra zdrowia. Krzywdzicie konkretne kobiety, konkretne osoby: matki, córki, wnuczki, siostry, żony i partnerki. Wypisywanie przez ten wyrok ze szpitala osób przed planowanymi legalnymi zabiegami przerywania ciąży z powodu ciężkich wad wrodzonych płodu to jest coś, co się dzieje obecnie w Polsce. To kobiety, które już nie otrzymają pomocy i będą zmuszone do porodów ciąż z wadami letalnymi, śmiertelnymi.

Krzywdzicie lekarki i pielęgniarki, które swoje siostry, córki, wnuczki, pacjentki będą musiały traktować w nieludzki i upokarzający sposób, odmawiając im opieki zdrowotnej. Bo teraz wszyscy lekarze i lekarki według was mają być Chazanami. To jest upadek moralny, krzywda kobiet i deptanie praw człowieka. Wykazywany na podstawie badań prenatalnych zespół Pataua czy zespół Edwardsa prowadzą do rozszczepu wargi i podniebienia, małogłowia, braku gałek ocznych. Do innych wad należy m.in. anencefalia, która charakteryzuje się brakiem lub szczątkowym rozwojem mózgowia, bezczaszkowiem. Syronmenelia polega na częściowym lub całkowitym zrośnięciu kończyn dolnych prowadzących do niedorozwoju pęcherza moczowego, niedorozwoju jelita. Ektopia serca polega na nieprawidłowym położeniu serca, które znajduje się poza obrębem klatki piersiowej. To tylko niektóre wady kwalifikujące do przerwania ciąży sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy go opublikujecie, kobiety będą musiały rodzić płody, rodzić dzieci, które rozwijają się z takimi wadami. Chciałabym usłyszeć od Ministerstwa Zdrowia, jakie dokładnie w 2019 r. były przesłanki przerywania ciąż. Niech kobiety wiedzą, na co je skazaliście. Niech wiedzą dokładnie, jakie były przesłanki. Chodzi o to, żeby mogły usłyszeć z waszych ust, na co chcecie je skazać, jakim torturom chcecie je poddać. Przez 9 miesięcy będą w ciąży, która skończy się tylko i wyłącznie cierpieniem i śmiercią. To są prawdziwe owoce waszej zbrodniczej, pomylonej ideologii. Ale żadna z kobiet nie będzie już szła sama. Będziemy je wspierać. Dlatego wnoszę również o informację, ile zabiegów przerywania ciąży odwołano od ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego o rozpoznaniach, w związku z którymi podejmowano decyzję o przerwaniu ciąży. Ile dzieci z zespołem Edwardsa i Pataua, bezczaszkowiem, kazaliście właśnie urodzić kobietom? Jak Ministerstwo Zdrowia ma zamiar przeorganizować publiczny system opieki zdrowotnej, złożony z podmiotów leczniczych podległych ministerstwu, aby w dobie pandemii koronawirusa, ale także w dobie barbarzyńskiego wyroku Trybunału Konstytucyjnego zapewnić efektywne wykonywanie świadczenia zdrowotnego w postaci przerywania ciąży zgodnie z ustawą z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, i to we wszystkich trzech przypadkach, do czasu opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a po jego opublikowaniu - w przypadku pozostałych dwóch przesłanek? Czy Ministerstwo Zdrowia ma zamiar, a jeśli tak, to kiedy i gdzie, ogłosić listę podmiotów leczniczych posiadających kontrakt z NFZ, których oddziały ginekologiczno-położnicze pozostają otwarte i przyjmują pacjentki w celu wykonania gwarantowanego świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w pkt 1? Ile z nich jest dostosowanych do potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami, o które podobno tak dbacie? Ile z tych gabinetów lekarskich, ile z tych szpitali położniczych jest dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Co zrobiliście od 2018 r. w sprawie dostępności gabinetów ginekologicznych? Tak dbacie o kobiety? Na wsi dostęp do gabinetów ginekologicznych praktycznie nie istnieje. Pora stanąć przed kobietami, które właśnie skrzywdziliście, i wytłumaczyć im wasze okrucieństwo. Siostry, nigdy nie będziecie szły same. Zawsze będziemy was wspierać. A ci, którzy chcą torturować kobiety, niech się z tego tłumaczą. Dziękuję serdecznie pani posłance.

Proszę bardzo.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Każdy obywatel naszego kraju ma prawo do życia, ma prawo do ochrony zdrowia, a to prawo ma mu zagwarantować władza publiczna.

Szanowni Państwo!

Te świadczenia winne być wykonywane na tych zasadach, jakie do tej pory były realizowane. Szanowni Państwo! Należy pamiętać o tym, że do tej pory również pracownicy ochrony zdrowia mieli możliwość korzystania z klauzuli sumienia.

Takie sytuacje się zdarzały, ale w takim przypadku osoby, które miały prawnie zagwarantowaną możliwość wykonania tego typu zabiegu, były informowane, gdzie te świadczenia mogą zostać wykonane.

Szanowni Państwo! Ta dostępność jest warunkowana wieloma czynnikami. Po pierwsze, jest to dostępność terytorialna. Tutaj dużą rolę odgrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, który kontraktuje świadczenia zdrowotne w różnych formach, w różnych rodzajach produktów i w różnej przestrzeni na terenie naszego kraju, analizując odpowiednie potrzeby zdrowotne. W ostatnim czasie, w ostatnich latach zwiększyliśmy ilość świadczeń udzielanych właśnie w ramach świadczeń z zakresu ginekologii i położnictwa. Po pierwsze, kontraktowane są świadczenia udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w ramach świadczeń z zakresu ginekologii i położnictwa, ale również w ramach świadczeń, które zostały wprowadzone przez ten rząd na podstawie ustawy „Za życiem”

Koordynowana opieka nad ciężarnymi jest realizowana na trzech etapach: na poziomie wojewódzkim, powiatowym oraz, przez ośrodek koordynujący, na poziomie ogólnopolskim. Tam właśnie kobiety, które dowiedziały się o problemach zdrowotnych dziecka poczętego, mogą uzyskać profesjonalną pomoc, mogą mieć wykonane badania, są otoczone opieką psychologiczną i psychiatryczną, której finansowanie według wskaźnika jest o 50% wyższe niż w pozostałych przypadkach. Te kobiety mają zabezpieczoną również możliwość wykonania badań prenatalnych. W Polsce mamy pięć ośrodków, które mogą udzielać pomocy dzieciom poczętym, u których stwierdzono wady. Te ośrodki przeprowadzają bardzo skomplikowane terapie, bardzo skomplikowane zabiegi operacyjne. Dzięki temu dzieci mają większą szansę na przeżycie.

Nie zapomnieliśmy również, realizując ustawę za życiem, o osobach, które zdecydowały się urodzić dziecko z problemami zdrowotnymi. Gwarantujemy im opiekę pediatryczną. Stworzono sieć dziecięcych ośrodków koordynujących, działających na poziomie poszczególnych województw, które opiekują się dziećmi, rodzinami -to jest problem całej rodziny - koordynując proces wspierania tych osób.

Nie zapomnieliśmy też o tych rodzinach, w których dzieci rodzą się z wadą letalną. Uruchomiliśmy sieć hospicjów perinatalnych, w których kobiety w ciąży, które noszą dziecko z wadą letalną, mogą liczyć na pomoc profesjonalistów, psychologów, psychiatrów. Takich hospicjów mamy w kraju 16. Ponad 500 tys. zł jest przeznaczane na opiekę właśnie w tym obszarze. Przede wszystkim chcemy jednak inwestować w zdrowie, stwarzać szanse na rozwój, na urodzenie zdrowego dziecka. Dlatego zależy nam na badaniach prenatalnych, które są realizowane i będą rozszerzane zgodnie z propozycją pana premiera Mateusza Morawieckiego.

Są to bardzo skomplikowane zabiegi, często kardiologiczne czy np. wykonywane u dzieci z przepukliną rdzeniowo-mózgową. To są zabiegi, które gwarantują dobrostan tych dzieci. Państwo pytacie, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o kadrę medyczną. Szanowni państwo, to za naszych czasów, już kilkakrotnie to mówiłam, zwiększyliśmy ilość uczelni medycznych, na których kształcimy lekarzy. Od 2015 r. powstało siedem nowych uczelni, które kształcą na wydziałach lekarskich. To daje średnio o 2 tys. więcej absolwentów niż było 6, 7 czy 8 lat temu. Proces kształcenia lekarza trwa długo, a specjalisty jeszcze dłużej. Dlatego borykamy się z problemem braku lekarzy. Zwiększamy ilość miejsc na studiach, zwiększamy ilość rezydentów. Z roku na rok ta liczba rośnie.

W związku z tym poszerzamy kompetencje położnych, które w dużej mierze przejmują opiekę nad kobietą ciężarną, realizują zadania wynikające z nowego standardu opieki okołoporodowej, który został przygotowany przez obecny rząd.

To my zapewniliśmy właśnie taką dostępność do świadczeń. Oczywiście wiemy, że jeszcze bardzo dużo przed nami. Wiele rzeczy jeszcze musimy udoskonalić, zmienić. Te działania są na bieżąco podejmowane. Ale podejmujemy działania, aby osoby potrzebujące wsparcia, kobiety z trudną ciążą, miały zagwarantowany dostęp do niego nawet w warunkach pandemicznych, aby miały dostęp nie tylko do lekarza ginekologa, położnej środowiskowej, lecz także do świadczeń specjalistycznych, bo one będą warunkowały dobrostan zarówno dziecka, jak i kobiety. Dziękuję bardzo, pani minister. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze zapisać się do głosu? To bardzo proszę. Proszę o zabranie głosu panią poseł Annę Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!

Pragnę przypomnieć, że perinatologia to specjalizacja, która pozwala leczyć matkę i pośrednio płód, ale także w przypadku różnych schorzeń bezpośrednich, bezpośrednio leczyć płód, o czym mówiła pani minister. Pragnę także zauważyć, że dzięki miniaturyzacji, dzięki ogromnemu postępowi w tzw. technice medycznej, dzięki takim aparatom jak USG, jak endoskopia możemy w życiu płodowym bardzo precyzyjnie leczyć dzieci. Chciałabym spytać o ten postęp na przestrzeni ostatnich lat. Ile już przeprowadzono operacji i w jakich bardzo skomplikowanych przypadkach możemy leczyć dziecko w życiu płodowym? Jakie polska medycyna, polska ginekologia ma w tym zakresie osiągnięcia?

Kończąc swoją wypowiedź, pragnę także spytać o bardzo ważną rzecz, związaną już z samymi badaniami prenatalnymi. Chodzi mi o wartość świadczeń zdrowotnych w tym zakresie w ostatnim roku rządów naszych poprzedników. Bardzo dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu panią poseł Monikę Rosę, Koalicja Obywatelska. Pani Minister! Wysoka Izbo! Aborcja w Polsce powinna być darmowa, legalna i bezpieczna, a dzięki edukacji seksualnej i dostępowi do antykoncepcji - także rzadka. Standardem krajów Unii Europejskiej jest dostęp kobiet do legalnej aborcji. Jest to kwestia praw człowieka, prawa do decydowania o sobie, prawa do bycia i życia na równi z innymi obywatelami, obywatelkami Unii Europejskiej. Ograniczenie prawa do aborcji to naruszenie prawa kobiet do życia, zdrowia, godności, prywatności, wolności od tortur i nieludzkiego traktowania. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale zakaz aborcji nie sprawi, że tych aborcji będzie mniej. Tych aborcji będzie tyle samo, tylko że poszukiwania drogi wyjścia z trudnej sytuacji dla kobiety będzie trudniejsze i doprowadzi to do wielu tragedii. Mam do pani minister pytania. Kiedy państwo rozszerzycie program badań prenatalnych? Teraz są przesłanki, które mówią o 35. roku życia albo o prawdopodobieństwie uszkodzenia płodu. Dlaczego nie wszystkie kobiety miałyby prawo skorzystać z tego programu? Poza tym chciałabym państwu powiedzieć, że kobiety z niepełnosprawnością fizyczną także zachodzą w ciążę, także uprawiają seks, natomiast dostęp do gabinetów ginekologicznych dostosowanych do potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami jest dramatycznie niski. Moje pytanie: Ile szpitali położniczych, ile gabinetów ginekologicznych jest dostosowanych do potrzeb kobiet z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym oczywiście fizycznymi?

Bardzo dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu panią poseł Wandę Nowicką, Lewica. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Za chwilę wejdzie w życie okrutne, nieludzkie, niehumanitarne prawo, które łamie w drastyczny sposób prawa kobiet, prawa połowy członków społeczeństwa, kobiet, które protestują na ulicach, a dzisiaj również strajkują poprzez odmowę świadczenia pracy. Prezes Kaczyński nie pozostawił żadnych złudzeń, nie ma żadnego współczucia, żadnej empatii dla kobiet. Prawo i Sprawiedliwość zdradziło kobiety, nie traktuje ich jak obywatelki, które mają prawo do życia, prawo do decydowania o swoim życiu prywatnym, prawo do godności i prawo do życia bez bycia torturowanym. To, co mówię, to nie jest tylko stanowisko posłanek i posłów opozycji czy kilkudziesięciu procent, 80%, społeczeństwa, które jest przeciwne temu drastycznemu prawu.

Mówią w nim: Polska zdecydowała się poświęcić prawa kobiet do bezpiecznej, legalnej aborcji z naruszeniem międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka. ONZ mówi: Solidaryzujemy się z kobietami w Polsce i ich dążeniami do równości. Wzywamy władze polskie do ochrony praw kobiet i mężczyzn, którzy protestują przeciwko temu.

Pokazują w sposób jednoznaczny, że prawa kobiet są prawami człowieka, a przez polski rząd, do którego ONZ apeluje, są łamane. I moje pytanie jest takie: Czy rząd zamierza wypowiedzieć wszystkie traktaty i konwencje międzynarodowe, które mówią o prawach kobiet, o prawie kobiet do samostanowienia o swoim życiu, o prawie do decydowania o swoim życiu i o wszystkich aspektach związanych z ciążą, macierzyństwem, porodem i własną płodnością? Czy to oznacza, że Polska w tej chwili stanie się.

Głos zabierze pan poseł Dariusz Klimczak, Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Szanowny Panie Marszałku! Chciałbym poruszyć dwa wątki. Pierwszy jest kontynuacją wystąpienia pani poseł Marceliny Zawiszy. Mianowicie chciałbym zapytać o wiejską drogę kobiety do ginekologa, jak ona dzisiaj wygląda, bo według ostatniej kontroli Najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie kobiety zamieszkałe na wsi miały utrudniony dostęp do ambulatoryjnych świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków publicznych. I choć standardy opieki okołoporodowej były jasno wyznaczone, część poradni ginekologicznych miała problemy z ich przestrzeganiem. Nie wszystkim kobietom w ciąży wykonano pełny zakres badań zalecanych standardami opieki okołoporodowej, wciąż też zdarzały się poradnie, które nie gwarantowały pacjentkom prawa do intymności. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia na koniec 2016 r. wynikało, że w wielu gminach wiejskich w ogóle nie było poradni ginekologiczno-położniczych, np. w moim województwie w 49% gmin, w co drugiej gminie. Pytanie: Jak dzisiaj wygląda dostępność do świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków publicznych na terenach wiejskich? Jakie są efekty wdrożenia zaleceń pokontrolnych NIK w aktualnej statystyce ministerstwa?

Chciałbym zapytać, ile w Polsce jest ośrodków diagnozy i terapii FAS, zespołu alkoholowego? Ile takich powstało i ile świadczy pomoc dla dzieci? Bardzo dziękuję. Chciałbym prosić o spokój na sali, niewymachiwanie palcem i niewykrzykiwanie „czas”, bo kiedy pani minister miała wydłużony czas o 5 minut, była także w taki sposób jak panie posłanki, które wydłużają swój czas, odpowiednio dobrze potraktowana. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja z kwarantanny.

W związku z tym postaram się jednak zadać pytania dość trudne, ale tej materii dotyczące. Pierwsza sprawa to dostępność do tych gabinetów. Pamiętajmy, że służba zdrowia, ta najbliżej pacjenta, czyli specjalistyczne gabinety lekarskie, pomijam szpitale, to jest dzisiaj inicjatywa prywatna, czyli to są po prostu prywatne poradnie, ośrodki. W związku z tym pytanie jest również do rządu, czy rząd rozmawiał chociażby z samorządowcami, żeby tam, gdzie istnieje rzeczywiście konieczność powołania takiej poradni, władze samorządowe również mogły w tym uczestniczyć, chociażby na poziomie czynszu czy najmu, by był zdecydowanie niższy, czy przez kwestie podatkowe, jakieś wspieranie tej działalności, ponieważ mają takie możliwości i takie prawo.

Czy w tej sprawie mamy jakieś pozytywne sygnały? Chciałbym usłyszeć, ilu rezydentów przygotowuje się do tej specjalizacji i kiedy należy się spodziewać zwiększonej liczby ginekologów i położników w polskiej ochronie zdrowia.

Czy są na to przeznaczone dodatkowe środki finansowe? Dziękuję bardzo. Życzymy zdrowia panu posłowi. Proszę o zabranie głosu panią poseł Zofię Czernow, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Kolejny obszar wykluczenia kobiet to brak opieki ginekologicznej nad kobietami z niepełnosprawnością. Tu jest prawdziwy dramat, proszę państwa. Kobiety z niepełnosprawnością bardzo rzadko korzystają z badań ginekologicznych, z profilaktyki.

Natomiast samotne kobiety niepełnosprawne mają wielkie problemy z badaniami. Z nich generalnie nie korzystają, i to zarówno z powodów logistycznych, ale też z powodów mentalnych i innych. Kobiety przebywające w ośrodkach, domach pomocy społecznej, innych ośrodkach, edukacyjnych również, młode dziewczyny - nie są objęte profilaktyką i badaniami kontrolnymi. To jest po prostu wykluczenie. I z jednej strony wynika to z braku dostosowania gabinetów ginekologicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale z drugiej strony nikt się tym nie zajmuje, nikt nie pomaga kobietom w dotarciu do takich badań. O badaniach prenatalnych wśród kobiet ciężarnych z niepełnosprawnością można zapomnieć. Ich po prostu nie ma i nikt się tym nie interesuje.

Jak wygląda to dotarcie? Pani minister Maląg bardzo cieszyła się wczoraj z opieki nad niepełnosprawnymi [[Dzwonek]] rodzinami. Ta opieka jest bardzo słaba, na najniższym poziomie w Europie. Kiedy ta sytuacja ulegnie zmianie? Proszę o zabranie głosu panią poseł Małgorzatę Prokop-Paczkowską, Lewica. Wysoka Izbo! Od czasu haniebnego wyroku pseudo-Trybunału Konstytucyjnego poszczególne frakcje obozu rządzącego próbują coś zrobić, aby się jakoś wyłgać, aby powiedzieć Polkom, że właściwie nic się nie stało. Jarosław Kaczyński wsadził na minę Kościół, który teraz kombinuje, jak się od was odciąć. Mateusz Morawiecki i Gowin próbują na swój sposób zamydlić kobietom oczy i mówić: na prawo aborcji to nie pozwalamy i nie pozwolimy, ale jak będziecie grzeczne. w swojej łaskawości może pozwolimy wam nie rodzić płodów bez głowy, serca czy mózgu. Polska prawica nie jest w stanie zaakceptować, że kobietom nie chodzi o pozwalanie im na to, co mają zrobić ze swoją ciążą.

Moje pytanie: Co rząd zrobi jeszcze, aby zrealizować swoje „nie pozwalamy” Gazowanie na ulicach już było. Zatrzymania są cały czas. Czy wprowadzicie godzinę policyjną przed piątkiem? Bo jak pewnie wiecie, będzie ogromny protest w piątek. Czy zatrudnicie na etatach bandziorów stadionowych, którzy nazywają się Strażą Narodową? Bardzo dziękuję.

Wysoka Izbo! Mam pytanie natury bardziej ogólnej. Otóż w lipcu br. kierownictwo Narodowego Funduszu Zdrowia zadeklarowało powołanie zespołu, którego celem miało być opracowanie planu przywracania pełnej dostępności świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a ograniczonych, jak wiemy, w wyniku pojawienia się pandemii koronawirusa. Zespół miał też rozeznać skalę ograniczeń w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej oraz dokonać oceny ryzyka związanego z przywracaniem pełnej dostępności tych świadczeń. Chciałbym zapytać: Czy taki zespół powstał, a jeśli tak, to czy znane są już wyniki jego działania? Zdrowia życzymy. Głos teraz zabierze pani poseł Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Panie i Panowie Posłowie! Chciałabym zacząć od kwestii pewnej hipokryzji całej prawicowej strony sceny politycznej, ponieważ zdajemy sobie sprawę z jednej rzeczy. Osoba zaradna, osoba zamożna nie będzie miała żadnego problemu z aborcją w Polsce, dlatego że do 9. tygodnia aborcja jest farmakologiczna i, szczerze mówiąc, zdobycie tego typu środków nie jest znowu tak trudne, jeżeli ktoś jest zaradny.

W związku z tym tak naprawdę ta zmiana doprowadza do sytuacji najbardziej tragicznej, bo wymaga pewnego heroizmu od kobiet. Nie każda musi być na to gotowa. I tak naprawdę nikt nikogo nie zmusza. Ktoś tutaj, słyszę czasem, roni krokodyle łzy nad kobietami, które biedne muszą dokonać aborcji, jak się potem będą czuły. To jest ich wybór. Chciałam spytać, jak to wygląda, ponieważ mam tu zestawienia dotyczące dwóch programów.

Proszę o zabranie głosu panią Katarzynę Kotulę, Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wady letalne to 80% przypadków legalnych zabiegów przerwania ciąży. Polska, szpital o III stopniu referencyjności. Płody umierają w kąciku noworodka i w inkubatorze. Owinięte w kocyk, czekają godzinami na śmierć. Nie stosuje się w stosunku do nich żadnych procedur medycznych, nie karmi, nie podaje środka znieczulającego. Położne i pielęgniarki czekają na ich śmierć. Płód czasem się dusi, umiera powoli, czasem kilka godzin. Bywa, że z głodu, przeważnie samotnie. Nie ma w Polsce jasnych przepisów, jak postąpić, a lekarze muszą rozstrzygać to sami, kierując się być może dobrem płodu, nakazami sumienia, religii, obawą przed posądzeniem o eutanazję. Reanimować? Podłączyć tlen? Chodzą słuchy, że niektórzy lekarze operują dla wprawy, która przyda się dla dzieci rokujących lepiej, a nie tych beznadziejnie. Jakie są procedury medyczne i wytyczne dotyczące postępowania w przypadku wad letalnych? I czy są one takie same jak te, które przytoczyłam w przykładzie ze szczecińskiego szpitala? Wiemy, że w Austrii podaje się środek znieczulający, fentanyl. W Polsce nie podaje się takich środków. Czy macie świadomość, że te płody umierają właśnie w ten sposób? Czy uważacie, że to jest etycznie moralne i humanitarne? Bo usta macie pełne frazesów o moralności i godności. Chciałabym też zapytać o procedury dotyczące kobiet. 2 miesiące temu w polskim szpitalu moja przyjaciółka, matka dwójki dzieci w piątym miesiącu ciąży dowiedziała się o tym, że płód nie ma wykształconego pęcherza i nerek. W momencie, w którym wywalczyła sobie prawo do aborcji, dostała do ręki tabletkę, dostała do ręki tekturowy basen. Polecono jej, aby udała się do łazienki, aby samotnie urodziła płód, nie patrzyła na ziemię i wezwała personel medyczny. To są te procedury, które obowiązują w Polsce. Chciałabym zapytać, czy takie są procedury (Dzwonek), czy to standard i czy to ma cokolwiek wspólnego z godnością, o której tyle mówicie, argumentując wyrok pseudotrybunału. To wy skazujecie te kobiety na takie cierpienie i pozbawiacie je godności i prawa wyboru. To wy pozbawiacie kobiety prawa wyboru. Dziękuję bardzo. Głos teraz zabierze pan poseł Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Jeszcze kilka lat temu, kiedy zajmowałem się opieką perinatalną w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, śmiertelność okołoporodowa dzieci była niezwykle wysoka, w szczególności wysoka w regionie, z którego pochodzę.

To pokazuje coraz lepszą, poprawiającą się opiekę okołoporodową dla kobiet w Polsce, lepszy sprzęt, programy profilaktyczne, dostępność opieki ginekologicznej, neonatologicznej, położniczej. Ale nadal - zawsze, bo zawsze może być lepiej - można zrobić więcej. I moje pytanie do pani minister jest takie: Jakie dalsze działania będą podejmowane, aby dalej poprawiać jakość opieki okołoporodowej? Bardzo dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu panią poseł Barbarę Nowacką, Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo! Tyle państwo mówicie o pomocy, a jak wygląda dostępność gabinetów ginekologicznych? Wygląda w ten sposób, że wiele kobiet do tych gabinetów dostać się nie ma jak, ponieważ, szczególnie w Polsce wschodniej i południowej, ta dostępność często oznacza kilkadziesiąt kilometrów. Gabinety czynne raz w tygodniu, na chwileczkę i wtedy nie ma jak.

Tak wam zależy na zdrowiu i życiu dzieci. No to co się stało z transplantologią dziecięcą? 509 dni czekają dzieci na zabieg transplantologii, zniszczonej notabene przez ministra Ziobrę w sposób okrutny i stricte polityczny. Transplantologia dziecięca w Polsce jest jedną z najgorszych i właściwie niefunkcjonujących. Dzieci umierają. W Internecie są zrzutki pieniędzy, żeby pomóc wyjechać rodzinom, które mają dzieci chociażby z chorobami kardiologicznymi, gdzieś za granicę i wykonać przeszczep, bo Polska tego nie świadczy, bo nie ma dobrych programów promocyjnych. Światowe Dni Transplantologii przecież były kilka dni temu, i co zrobił polski rząd, w jaki sposób zajmuje się tym? Klinika w Krakowie, też zajmująca się transplantologią, przecież zamknięta. Szanowni Państwo! Jeżeli chcecie realnie pomagać, to pomóżcie tam, gdzie trzeba pomóc biednym i wykluczonym, gdzie trzeba pomóc chorym, a przestańcie uprawiać ideologię i toczyć wojnę z kobietami. Dajcie kobietom wybór. Kobiety wybiorą mądrze, ale dajcie też narzędzia, szpital i opiekę zdrowotną. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią poseł Katarzynę Kretkowską, Lewica. Wysoka Izbo! Wybór to nie nakaz, jak pada wielokrotnie z tej trybuny. W krajach, w których jest dostęp do wyboru, jest mniej zabiegów przerywania ciąży niż w krajach, gdzie ten wybór jest zakazany. O tym wszyscy wiemy, ale państwo z PiS udajecie, że o tym nie wiecie. I udajecie, że nie wiecie o tym, że od czasu, gdy ograniczono dostęp do aborcji, wykonano w Polsce ponad 4 mln tych zabiegów. Mam pytania dotyczące dostępu i do badań prenatalnych, i do badań prenatalnych po tym, jak ten wyrok pseudotrybunału wejdzie w życie. Tutaj bardzo dużo słyszeliśmy pięknych słów od pani minister. Ja chciałem zarówno panią poseł, jak i panie posłanki prosić o umożliwienie dokończenia wystąpienia koleżance. Jak rząd zamierza przeciwdziałać odmowie wykonywania badań prenatalnych przez publiczne placówki ochrony zdrowia, gdy te placówki będą się obawiały zarzutu, że zamierzają podżegać do nielegalnych zabiegów przerywania ciąży, gdy te badania wykażą letalną wadę płodu? Jak zamierzacie temu przeciwdziałać? W placówkach publicznych, czy to w prywatnych z podpisaną umową z NFZ, czy w publicznych szpitalach, nie powinni być zatrudniani lekarze, którzy chcą się kierować klauzulą sumienia i odmawiać zabiegów przewidzianych prawem, dlatego że to nie zgadza się z ich sumieniem. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby lekarze, którzy kierują się klauzulą sumienia, funkcjonowali w katolickich placówkach ochrony zdrowia (Dzwonek), ale publiczne placówki ochrony zdrowia nie powinny takich ludzi zatrudniać.

Ile badań i ile środków przewiduje się, o tym mówiła pani minister, na przyszły rok na badania prenatalne? Ile szczególnie będzie tych badań wykonywanych w Wielkopolsce? Jeszcze ostatnia uwaga. Państwo mówicie pięknie o hospicjach perinatalnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby katoliczki czy osoby, które decydują się urodzić, korzystały z tych hospicjów. Ale to nie może być tak, że zmuszacie kobiety do korzystania z tych hospicjów. Kobiety, które nie chcą rodzić dziecka, które będzie w cierpieniu umierać, powinny mieć dostęp do zabiegu przerwania tej ciąży. Proszę bardzo panią poseł Barbarę Bartuś, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Naszej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy zasadniczej.

Szanowni Państwo! Droga Opozycjo! Totalna Opozycjo! Zostaliście wybrani do polskiego Sejmu, żeby reprezentować Polki i Polaków, a robicie nam wszystkim piekło. Wyprowadzacie ludzi, młodych ludzi na ulice, pod fałszywymi hasłami. W imię tak zwanej legalnej aborcji? Czy was interesują cokolwiek te młode kobiety, które kiedyś będą podejmować może świadomą może nieświadomą decyzję o tym, że mogą zostać matkami? Ja jestem ze wsi, ja wiem, jaki miałam dostęp do lekarza ginekologa, gdy ja byłam w ciąży. Wiem to i wszystkie te troski, obawy, rozumiem. I nad tym powinniśmy pracować - żeby pomóc, żeby pomóc, a nie namawiać do przestępstwa, do szukania wyjazdów za granicę. To co znaczy, że będziemy za chwilę mówić, że ci, którzy są bogatsi, mają lepszy dostęp do płatnego zabójcy niż ci, którzy są biedniejsi, bo ich na to nie stać? Są poważne problemy, są problemy, które się pojawiają w ciąży. Ale też mamy inne problemy. Przecież może być zdrowa ciąża (Dzwonek), a dziecko urodzić się z porażeniem mózgowym. Jest wiele, wiele problemów. Oczywiście, że to wszystko jest za mało. Ostatnio usłyszałam, że jest problem z dostępem do rehabilitacji ruchowej, właśnie dla dzieci. Czy są jakieś ograniczenia, limity, kiedy mamy pełną niepełnosprawność? Czy te kobiety, te rodziny mogłyby uzyskiwać większą pomoc? Tu, dzisiaj, szczególnie teraz, w okresie pandemii. Nie wyprowadzać młodych i nie tylko młodych na niebezpieczeństwo na ulicy. Bardzo dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu panią poseł Iwonę Marię Kozłowską, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pani minister tak pięknie mówiła o dostępie kobiet do gabinetów ginekologicznych, o wspaniałych badaniach, które idą z duchem nowoczesności. O tym, że każda kobieta może chronić swoje życie i życie i zdrowie swojego dziecka.

78% kobiet nie robi podstawowych badań w okresie ciąży, które zaleca lekarz. 20% kobiet nie ma nawet dokumentacji przebiegu ciąży. Więc jak to wygląda, jeżeli chodzi o dostępność gabinetów ginekologicznych, badań, opieki i wsparcia lekarzy ginekologów dla kobiet na wsiach? I bardzo proszę o przygotowanie na piśmie informacji, jaka jest dostępność przychodni i gabinetów ginekologicznych na wsiach w województwie kujawsko-pomorskim.

Ale pewnie jak otrzymam od pani na piśmie informację, to będę to wiedziała i będę znała wszystkie szczegóły. Moje kolejne pytanie dotyczy praktycznych skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a pytanie kieruję do sygnatariuszy tego wniosku. Kanwa praktyczna. Kobieta zachodzi w bliźniaczą ciążę.

W związku z tym rodzice - katolicy, głęboko wierzący - podejmują wraz z lekarzami decyzję o usunięciu płodu. Szanowni państwo, urodziło się zdrowe maleństwo, jest szczęśliwa rodzina.

Bardzo dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu panią poseł Monikę Falej, Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiaj tylko 9% szpitali w Polsce wykonuje zabiegi legalnej aborcji pomimo podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prawo do przerywania ciąży jest zagwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, jako dostęp do świadczeń medycznych. Aborcja to zabieg medyczny, jak każdy inny.

Przecież to nie jest tak, że wady letalne nie występują na Podkarpaciu. Kobiety z tego regionu albo jadą za granicę, albo dokonują zabiegu w klinice, biorąc kredyt, bo Polska odmawia im tego prawa, które im przysługuje. Czy macie świadomość, że będziecie wspierać podziemie aborcyjne w Polsce oraz turystykę aborcyjną? Aborcja była, jest i będzie, tylko w jakich warunkach i za jaką cenę? Dlaczego skazujecie kobiety na tortury i popadanie w zadłużenie? Bo ważniejsza jest klauzula sumienia i fanatyzm religijny? Pięknie pani minister mówiła też o dostępności lekarzy ginekologów, gabinetów ginekologicznych, w tym dla kobiet z niepełnosprawnościami. Dlatego zwracam się z prośbą o informację, ile gabinetów w województwie warmińsko-mazurskim jest przystosowanych do osób z niepełnosprawnością. Proszę o informację, ile kobiet z niepełnosprawnością z tych gabinetów skorzystało. Dziękuję bardzo. Nie będziesz szła sama. Te informacje poproszę oczywiście na piśmie. Bardzo dziękuję. Witam serdecznie. Panie marszałku, czy jestem słyszany? Tak, proszę bardzo. Witam serdecznie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Myślę, że w tej debacie niepotrzebnie pojawiły się emocje, duże emocje.

Trzeba powiedzieć, że nieprawdą są kwestie związane z pogorszeniem dostępu do gabinetów ginekologicznych dla kobiet na wsi, bo to za naszych rządów poluzowano pewne twarde kryteria, które wprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia, a gabinety - przypomnę - są prywatne i są otwierane w różnych małych miasteczkach, na wsi, w innych miejscach przez określonych lekarzy, i to oni powinni dbać również o zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Po pierwsze, transplantologia. To nie jest tak. Muszą być dawcy, aby tę transplantację móc przeprowadzić. W Polsce jesteśmy gotowi do transplantacji. Wreszcie muszę zaprotestować w imieniu wszystkich lekarzy. Nie może być tak, i tak nie jest, pani poseł, że ktoś operuje, dokonuje eksperymentów na dziecku, które było poddane aborcji, które nie ma prawa do życia. Nic takiego w Polsce nie ma miejsca i to jest skandal, że ktoś o coś takiego lekarzy oskarża. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu panią poseł Anitę Kucharską-Dziedzic. Przepraszam bardzo, ale była umowa, że. Wysoka Izbo! Pani Bartuś powiedziała, że młode kobiety będą podejmować decyzję świadomie lub nieświadomie. To jest clou sporu o legalność aborcji - żeby wszystkie kobiety podejmowały te decyzje świadomie, zawsze świadomie i zawsze samodzielnie i żeby nikt im się w te decyzje nie wtrącał ani nie odbierał podmiotowości ludzkiej. Bo czy jest to podmiotowość świecka, czy religijna, to nie ma żadnego znaczenia, bo i świeccy, i religijni ludzie mają wolną wolę i są podmiotami, a nie przedmiotami. Ale rozumiem, że pani poseł w zdenerwowaniu powiedziała coś, czego tak naprawdę nie chciała powiedzieć. To wyraz strachu, strachu o to, że na ulicach jest w tej chwili niewiele kobiet w wieku menopauzalnym czy panów w andropauzie. Na ulicach są przede wszystkim ci młodzi ludzie, którzy chcą podejmować decyzje dotyczące swojej płodności i rodzicielstwa samodzielnie i świadomie. To są ich decyzje związane z ich życiem. Nie chcą, żeby ktokolwiek im się w te decyzje wtrącał.

To jest, proszę państwa, państwowy protekcjonalizm podszyty moralizatorstwem, dzielenie kobiet na te, którym pozwoli się terminować ciążę, i te, którym się zabroni. Zdrowie psychiczne jest mniej ważne. Możesz się zabić, trudno. Państwo ci pozwoli terminować ciążę, jak masz raka. Czy ta ciąża, którą donosisz, spowoduje, że nigdy już nie urodzisz? O, jaka szkoda. Ale widocznie Bóg tak chciał.

Dziękuję bardzo. Czy koledzy z Koalicji Obywatelskiej coś uzgodnili? Pan poseł Szczerba teraz zabiera głos?

Panie marszałku, dziękuję. Szanowni Państwo! Poseł Latos mnie doskonale zna. To jest kolejny poseł, który dostał postulaty, z którymi spotykałam się nawet w różnych audycjach radiowych, i zna problemy środowiska osób z niepełnosprawnościami. To jest poseł, który wie, jak wygląda nasze realne życie. Natomiast to, co się wydarzyło przed chwilą. Państwo z PiS nie wiecie, co macie zrobić z tym bałaganem, z tym, co teraz robicie. Bardzo proszę, żeby nie mieszać do tego wszystkiego naszych dzieci, niepełnosprawnych, już po 18. roku życia.

Przecież nie dajecie nam pomocy. Nie ma asystentów, nie ma turnusów rehabilitacyjnych, co chwilę to powtarzam, a panie co chwilę krzyczą na mnie, że mówię nieprawdę. Mówię prawdę. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią poseł Agnieszkę Soin, Prawo i Sprawiedliwość.

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Pani Minister! Wysoka Izbo! Wcześniejsze wykrycie zaburzeń płodu możliwe jest m.in. dzięki badaniom prenatalnym, które wykonane na odpowiednio wczesnym etapie ciąży umożliwiają rozpoczęcie leczenia już w łonie matki. Obecnie refundowane są badania prenatalne dla grupy kobiet, które mają wskazanie do ich wykonania.

Bardzo dziękuję. Pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz, Koalicja Obywatelska, zabierze głos. Panie Marszałku! Nie mam wątpliwości co do tego, że kobiety powinny mieć zagwarantowane prawo wyboru, ale mam do pań pytanie: Czy panie w ogóle sobie zdają sprawę z tego, jakie konsekwencje wywoła wprowadzenie w życie tego waszego bestialskiego prawa zakazującego usuwania ciężko chorego, uszkodzonego płodu? Prof. Matyja, szef Naczelnej Izby Lekarskiej, powiedział bardzo jasno: „Praktycznie badania prenatalne będą niepotrzebne. Bo skoro one nie prowadzą do niczego, to tylko byłyby elementem badań naukowych” Czy panie sobie zdają sprawę z tego, jak wiele tak bardzo potrzebnych badań, tak bardzo potrzebnych terapii nie zostanie przeprowadzonych ze względu na wprowadzane przez państwa barbarzyńskie prawo? Jaki będzie praktyczny efekt tych bestialskich przepisów, tego prawa, które zostało wprowadzone w życie, właśnie ze względu na efekt mrożący, który ten barbarzyński nakaz wywoła? Do ilu dramatów to doprowadzi? Do jak olbrzymiego cierpienia? Ile dzieci przez was straci szansę na skuteczne leczenie prenatalne? Sama, kiedy byłam w ciąży i drżałam o zdrowie swojego dziecka, chciałam wykonać badanie prenatalne i odmówiono mi tego badania, mówiąc wprost: Po co ono pani? Co pani zrobi z takim wynikiem? Lekarka powołała się na klauzulę sumienia. Zmieniłam lekarza, ale historia miała dalszy ciąg. W 20. tygodni mojej ciąży wykryto u mojego synka na szczęście później niepotwierdzone schorzenie, które musiałoby zostać zoperowane w ciągu kilkudziesięciu godzin po porodzie, co oznaczało, że nie będę mogła rodzić w lokalnym, powiatowym szpitalu, tylko w specjalistycznej klinice. Bez badań prenatalnych, które właśnie zamroziliście, nawet nie miałabym takiej wiedzy. Ja nie miałabym takiej wiedzy, a moje dziecko nie miałoby szansy na życie w zdrowiu. Nie miałabym szansy nawet zawalczyć o zdrowie swojego dziecka, bo jakaś religijna fanatyczka chciała mnie tego prawa pozbawić, powiedziała: Niepotrzebne są pani badania prenatalne. Żadna matka, żaden ojciec wam nie daruje, jeżeli faktycznym skutkiem tego zakazu będzie niewykonywanie badań prenatalnych. Dziękuję bardzo.

Pani Minister! Wysoka Izbo!

Pani poseł Zawisza przedstawiła przerażający leksykon chorób bardziej lub mniej przerażających, również rozszczepienie wargi. Czy prawdą jest, pani minister, że większość aborcji, które w ostatnich latach zostały wykonane, wykonano z powodu podejrzenia u dzieci trisomii, czyli zespołu Downa? Mam również apel do pań po lewej stronie, ubranych tak żałobnie, żeby nie używały słów, których znaczenia nie rozumieją. Proszę państwa, barbarzyńca to osoba, która nie korzysta z dorobku swojej cywilizacji, a naszym dorobkiem cywilizacyjnym jest niezabijanie dzieci, również dzieci niepełnosprawnych. Humanitarny, czyli mający na celu dobro człowieka, poszanowanie jego praw.

Czy mam ogłosić przerwę, czy kontynuujemy? Proszę bardzo, głos teraz zabierze pan poseł Michał Gramatyka. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Historia prawdziwa, mój bliski przyjaciel jest ginekologiem. Pani Joanna, lat 29, pierwsza ciąża, 10. tydzień. Obraz USG pokazuje nieprawidłową budowę płodu, podejrzenie defektu głowy.

Dzisiaj badania prenatalne, o które tutaj tyle sporów już było, w szczególnych przypadkach są refundowane. Pytanie: Czy po tym tzw. wyroku są państwo w stanie zagwarantować, że ta refundacja pozostanie, że nikt nie wpadnie na pomysł, żeby ją zabrać i tym samym pozbawić kobiety możliwości przeprowadzenia badań prenatalnych? Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Pawła Rychlika, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo!

Będę zalecał wprowadzenie badań prenatalnych dla wszystkich, nie tylko dla kobiet powyżej 35. roku życia. czy z powikłaniami ciąży, żeby jak najwcześniej rozpoznać rozwój życia. To słowa pana premiera Mateusza Morawieckiego odnośnie do wypowiedzi pani poseł Gasiuk-Pihowicz, ale jej już na sali nie ma po odegraniu teatru. Pani Minister! Dostępność świadczeń to przede wszystkim wiedza o możliwości skorzystania z takiej opieki. Bazując na braku świadomości, jeśli chodzi o pewne zagadnienia, w przestrzeni publicznej, a także niestety wśród niektórych posłów, co dzisiaj dobitnie widzimy, chcę zapytać: W jaki sposób hospicja perinatalne wpływają na opiekę nad kobietami ciężarnymi? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Głos teraz zabierze pani poseł Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo się cieszę, że po wczorajszym bezpodstawnym wykluczeniu mogę dzisiaj z powrotem reprezentować swoich wyborców i swoje wyborczynie. Od tygodnia kraj żyje protestami. Po pseudowyroku TK zdezorientowani są także ginekolodzy i ich pacjentki, które nie wiedzą, czy zdążą zadecydować o swoim zdrowiu, ciele, a nawet o całym dalszym życiu swojej rodziny. Lekarze nie wiedzą, czy mogą leczyć i ratować życie pacjentek i czy za to nie skończą w więzieniu. W imieniu ginekologów, kobiet i całej protestującej ulicy pytam dzisiaj rząd PiS-u: Dlaczego tak okrutnie znęcacie się nad polskimi rodzinami? W imię utrzymania władzy jednej partii? Jako posłanki od tygodnia chodzimy na ulicę łagodzić konflikty, mediować, rozmawiać z policjantami i protestującymi, by nie polała się polska krew, a czasem jest naprawdę gorąco, bo pękają nerwy po obu stronach. Raz się uda, a raz nie, ale robimy, co możemy, mediujemy. A teraz inny poseł, poseł Kaczyński, w dodatku odpowiedzialny za obronność i bezpieczeństwo, wzywa do wojny domowej i obrony partyjnych interesów, bo przecież kościoły to przybudówki partii PiS, tam nie ma Boga, tam jest twarda polityka i kasa, do tego doprowadziliście. Pośle Kaczyński! Był pan chociaż raz przez ostatni tydzień porozmawiać z kobietami, zapytać, czego oczekują, dlaczego wychodzą na ulice? Bo byłam trzy razy pod pana domem i jakoś pana nie widziałam. Kryje się pan za kordonem policji, za ochroniarzami za nasze pieniądze. Ma pan coś do powiedzenia narodowi, to proszę wyjść na ulicę i powiedzieć to kobietom prosto w twarz. Każda dyktatura kiedyś upadnie. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią poseł Joannę Borowiak.

Na tym kończymy. Wysoki Sejmie! Do posłów totalnej opozycji: nie kłamcie, przestańcie kłamać. To nie jest prawda, że chodzicie na marsze po to, żeby uspokajać osoby, które tam są. Robicie sobie sweet focie tylko po to, żeby zaistnieć w mediach społecznościowych. A teraz przechodzę do informacji bieżącej. Obowiązkiem państwa jest roztaczanie opieki nad kobietami, które spodziewają się dziecka. Zadania w tym zakresie realizuje wprowadzona w 2006 r. opieka koordynowana nad kobietą w ciąży.

Pani Minister! Mam pytanie. W jakiej wysokości środki finansowe wydatkowano na tę formę wsparcia kobiet? Bardzo dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu panią poseł Monikę Wielichowską, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Wprowadziliście recepty na pigułkę dzień po, choć w większości krajów Unii Europejskiej jest ona dostępna bez recepty. Ratyfikowana konwencja o zwalczaniu przemocy wobec kobiet to niezrealizowany dokument, który wielokrotnie chcieliście wypowiedzieć. Uderzacie w organizacje kobiece, które kobietom pomagają, które kobiety wspierają, którym kobiety ufają. Klauzula sumienia ma się dobrze. Ministerstwo Zdrowia w reklamówkach zachęca do rozmnażania (Dzwonek) się jak króliki. Kiedy pod waszymi rządami Polska staje się ciemnogrodem, kiedy dostęp do medycyny XXI w. zastępujecie ideologią, kiedy z buciorami wchodzicie w życie, wybory, decyzje i wolności kobiet, zabierając im możliwości decydowania o sobie, posłanki PiS ubierają się na biało, a premier mówi: Będę zalecał wprowadzenie badań prenatalnych dla wszystkich kobiet. Jak to zrobicie? Kiedy? Jak? Gdzie? Za co? Jak to zrobicie? Czy ma pani świadomość, że w niektórych województwach nawet 70% gmin nie ma gabinetu ginekologicznego? Kobiety nie mają dostępu do gabinetu ginekologicznego. Tym się najpierw zajmijcie, dostępem do ginekologa, do możliwości zrobienia cytologii. Tym się najpierw zajmijcie, zamiast podpalać, podżegać i dolewać benzyny do obywatelskich protestów, wyręczać się pseudo-Trybunałem Konstytucyjnym i napuszczać ludzi na siebie. Kaczyński dobrze wiedział, że kobiety nie oddadzą swoich praw i wolności walkowerem. Wiedział, a pomimo to cynicznie to zrobił. To niebywałe, to niewybaczalne, to skrajnie odpowiedzialne. Proszę o zabranie głosu pana posła Jakuba Rutnickiego, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dlaczego protestują? One walczą o własną godność. One walczą o prawo do samostanowienia. Ale właśnie tą postawą, którą wy reprezentujecie, tą sytuacją, za którą odpowiedzialny jest Jarosław Kaczyński i jego odkrycie towarzyskie, pani Przyłębska, doprowadzicie do katastrofy demograficznej.

Wykorzystujecie go tylko dlatego, że nie radzicie sobie z pandemią. Spójrzcie na to w perspektywie kilku czy kilkunastu lat. Młode Polki walczą o swoje prawa, młode Polki protestują dlatego, że chcą w spokoju zachodzić w ciążę i rodzić dzieci. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią poseł Teresę Wargocką, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Informacja bieżąca złożona przez Lewicę, przez Platformę faktycznie miała być wyrazem troski o zdrowie kobiet w ciąży - liczba lekarzy, gabinetów ginekologicznych dla osób niepełnosprawnych, badania prenatalne.

Dokładnie to samo. Prawo do życia człowieka jest prawem najwyższym. Nie można prawa do życia porównywać z innymi prawami i stopniować. Prawo do życia człowieka wynika z jego godności, jaką mają wszyscy ludzie. I Trybunał Konstytucyjny nie mógł inaczej orzec, państwo dobrze wiecie. Gdybyście byli uczciwi i chcieli powiedzieć kobietom w Polsce, co oznacza wykreślenie z ustawy przesłanki eugenicznej, byście powiedzieli im prawdę. Jeżeli jesteś w ciąży powikłanej, jeżeli twoje dziecko może być chore, niepełnosprawne, prawo do życia osoby niepełnosprawnej nie jest różnicowane, czy jesteś człowiekiem dorosłym, czy jesteś człowiekiem w łonie matki - to mówi prawo. Dlaczego jest taki krzyk? W Polsce nigdy nie było prawa do aborcji. Była ustawa o ochronie i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, tych trzech. Jeżeli życie kobiety jest zagrożone, lekarz ma obowiązek ratować kobietę. Nadal ciąża z gwałtu jest przesłanką do tego, żeby ten problem został rozwiązany. Bardzo proszę, nie kłamcie, nie manipulujcie. Jeżeli mówicie młodzieży na swoich bluzkach, że aborcja jest okej, to ja współczuję tej młodzieży, zmanipulowanej, zniszczonej moralnie, tym młodym dziewczętom, które będą miały lęk przed macierzyństwem. To jest pokolenie, które było wychowane przez liberalną lewicową władzę: róbta, co chceta. Dziękuję bardzo. Na tym listę osób zapisanych do dyskusji wyczerpiemy. Będzie miała czas pani posłanka przedstawicielka wnioskodawców. Panią minister będziemy prosili tym razem o reżim czasowy - 5 minut. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 27 lat temu. Jarosław Kaczyński podniósł rękę za kompromisem aborcyjnym. W sytuacji, w której mamy do czynienia z ciężkim, nieodwracalnym uszkodzeniem płodu, kobieta może decydować. Jarosław Kaczyński mówi polskim kobietom, że to on będzie decydował, a nie one w sytuacjach dramatycznych, sytuacjach traumatycznych, w sytuacjach, które są psychicznymi torturami. Nie ma nic bardziej niegodnego niż te głosy, które płyną z tej strony sali. Szanowne panie posłanki i panowie posłowie z PiS, dziecko z bezmózgowiem, dziecko z bezczaszkowiem, dziecko bez ukształtowanych organów nie jest dzieckiem z niepełnosprawnością.

Szanowni Państwo! Mówicie o badaniach prenatalnych. Konsultant krajowy do spraw perinatologii prof. Mirosław Wielgoś mówi: Część ginekologów będzie unikać diagnostyki prenatalnej. Lekarze będą się obawiać, że w razie powikłań zostaną posądzeni o celowe działanie i pociągnięcie do odpowiedzialności. Pan premier mówi, że będzie rozwijał diagnostykę prenatalną, a konsultant krajowy pani minister i pana ministra mówi, że to jest tak naprawdę cofanie tej dyscypliny medycznej. Naprawdę opanujcie się. Dzisiaj zadaniem nas wszystkich jest stanąć przy polskich kobietach. Prosimy pana posła Tomasza Latosa o wygłoszenie sprostowania. Jestem słyszany, tak? Tak. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie powiedziałem ani jednego słowa, które było mi przypisane. Gorąca prośba. Słuchajmy siebie uważnie, cytujmy precyzyjnie. Ja nic takiego, co było mi zarzucane, nie powiedziałem. Przy okazji chciałbym wyrazić szacunek wobec wszystkich osób niepełnosprawnych. Kłaniam się. Proszę panią poseł Marcelinę Zawiszę jako przedstawicielkę wnioskodawców o zabranie głosu. Jeszcze raz ponawiam prośbę o zachowanie reżimu czasowego. Mamy na wypowiedź 5 minut. Pozostałe kwestie proszę przekazać posłom na piśmie. Wysoka Izbo! Szkoda, że nie będę miała możliwości ustosunkowania się do wielu państwa wypowiedzi, ponieważ one w wielu przypadkach mijają się z prawdą, a wręcz są nieprawdą. Na początek chciałabym jednak mimo wszystko stanąć w obronie lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Mamy wspaniałych lekarzy, którzy zrobią wszystko, aby w tych trudnych momentach zapewnić komfort zarówno rodzącym, jak i małym dzieciom. Szanowni Państwo! Wskaźniki mówią za siebie.

Badania prenatalne są w Polsce realizowane w coraz większej ilości, z roku na rok przeznaczamy coraz większe kwoty.

Skorzystało ponad 126 tys. matek.

Pani poseł Porowska pytała, w jaki sposób zwiększa się ilość badań USG. W 2015 r. było 121 tys., w tej chwili mamy 162 tys. Zwiększamy ilość badań i będziemy zwiększać, dlatego że one są potrzebne m.in. po to, abyśmy mogli w sposób profesjonalny pomagać tym dzieciom, abyśmy mogli wykonywać zabiegi, które są możliwe i dostępne w naszym kraju, a w wielu krajach Unii Europejskiej i na świecie są niedostępne. To są zabiegi kardiologiczne, zabiegi na nerkach, zabiegi dotyczące układu nerwowego.

A więc jeszcze raz państwu podam konkretne dane z 2019 r. Jeżeli chodzi o aborcje wykonane z powodu trisomii chromosomu 21 bez współistniejących wad, było to 271 przypadków, a ze współistniejącymi wadami somatycznymi - 164. To są, proszę państwa, zespoły Downa, czyli ponad 430 na 1074 to były aborcje dzieci, które posiadały wadę genetyczną zespołu Downa.

Poza tym jedna z pań poseł twierdziła, że w wielu województwach nie ma możliwości wykonania tego typu zabiegów.

Szanowni państwo, wielu z państwa pytało też i podawało dane, które są niezgodne z prawdą, np. że liczba zabiegów transplantacji u dzieci i młodzieży spada. Jest to nieprawda, proszę państwa. W tym roku dokonaliśmy więcej przeszczepów, np. serca, niż w roku 2015. Te dane są dostępne i możemy państwu je dokładnie pokazać.

Z roku na rok wydajemy coraz więcej środków na badania, na opiekę prenatalną i opiekę koordynowaną. Stworzyliśmy nowy produkt: koordynowana opieka nad ciężarnymi. Ona gwarantuje właśnie specjalistyczną opiekę kobietom, u których zdiagnozowano ciążę z problemami zdrowotnymi. To właśnie w ośrodkach specjalistycznych, na poziomie województw, są ośrodki koordynujące - tam jest prowadzenie takiej ciąży plus tam może się odbyć rozwiązanie takiej ciąży i tam też jest zabezpieczona opieka hospicyjna czy paliatywna, jeżeli jest wymagana. Od tego są te ośrodki. Koordynowana opieka nad ciężarnymi w tej chwili jest finansowana dodatkowo, bezlimitowo, ponad 350 mln zł wydajemy rokrocznie na finansowanie tych świadczeń. Było pytanie dotyczące ośrodków zajmujących się leczeniem FAS. I jeszcze jedno - wsparcie psychiczne i psychiatryczne. Na początku wypowiedzi to mówiłam. Kobiety, u których zdiagnozowano trudną ciążę, mają zapewnioną opiekę psychologiczną i psychiatryczną i te świadczenia są finansowane wskaźnikiem (...) dodatkowo 50%. Czyli tak naprawdę w interesie świadczeniodawcy jest przyjmować te kobiety po to, aby im zapewnić tę opiekę. Kwestia dostępności świadczeń. Szanowni państwo, pamiętajmy o tym, że zmieniliśmy system organizacji ochrony zdrowia. Wiele szpitali w Polsce w ryczałtach posiada środki finansowe na poradnie ginekologiczno-położnicze dla

poszczególnych województwach, to zgodnie z państwa życzeniem odpowiemy na piśmie. Wypowiedź ta kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego.

Obecnie przystąpimy do stwierdzenia kworum. Proszę o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu.

Stwierdzam, że mamy kworum. Mam zgłoszenia wniosków formalnych. Bardzo proszę, z pierwszym wnioskiem pan poseł Cezary Tomczyk, klub Koalicji Obywatelskiej. 1 minuta, panie pośle. Wysoka Izbo! Wnoszę o rozszerzenie porządku dziennego o raport o stanie bezpieczeństwa państwa. To pan, panie premierze, odpowiada dzisiaj za bezpieczeństwo w Polsce. Wczoraj wzywał pan do samosądów, do budowania PiS-owskich bojówek, które mają być wysyłane przeciwko. Pan wczoraj wystąpił przeciwko. Wprowadza pan opinię publiczną w błąd. To jest nie tylko głęboko niemoralne, nie tylko skandaliczne, ale jest to ciężkie przestępstwo przeciwko narodowi i przeciwko polskim obywatelom. Ciężkie przestępstwo, za które będzie pan musiał zapłacić. Wypuszczacie prowokatorów przeciwko protestującym. Agenci ABW wjeżdżają w tłumy protestujących, nie ma żadnych zarzutów. Jednocześnie wykorzystujecie sytuację, chcecie stawiać zarzuty posłom opozycji? Za to, że walczą z telewizją publiczną? Że chcą prawdy w Polsce? Tak, chcemy prawdy w Polsce, żądamy prawdy o epidemii. Żądamy prawdy w telewizji publicznej, tu, natychmiast. Tu, panie premierze, bo pan za to bezpośrednio odpowiada, za to, co dzieje się w Polsce, to jest pana odpowiedzialność i pana krew na rękach.

W trybie takim, że członkowie rządu mają prawo zabierać głos w każdym momencie.

Wysoka Izbo! Tu padło szereg kłamliwych zarzutów, i to na zasadzie takiego całkowitego odwrócenia się od prawdy. Mamy dzisiaj w Polsce, Wysoka Izbo, bardzo wysoki stan zagrożenia z powodu epidemii. To państwo twierdzą, że nie słyszycie, wobec tego mówię bez maseczki. Otóż ten stan wyklucza (Dzwonek) jakiekolwiek spotkania publiczne powyżej pięciu osób. Odbywają się z waszego podjudzenia. setki i tysiące różnego rodzaju demonstracji. A jednocześnie głosicie idiotyczne. No, może mnie pani obrażać, ale nie jest pani w stanie.

Panie Nitras, ostrzegam pana.

Wy w tej chwili w imię własnych interesów, małych, brudnych interesów, interesów Nowaka, [[Oklaski]] wy w imię tych interesów rozwalacie Polskę, narażacie na śmierć mnóstwo ludzi. Jesteście przestępcami. Jesteście przestępcami. Jest przestępstwo spowodowania niebezpieczeństwa powszechnego. Wy, wzywając do demonstracji, powodujecie tego rodzaju niebezpieczeństwa.

Na końcu, po tym wystąpieniu, po wnioskach formalnych udzielę panu głosu. Ale proszę tylko w trybie sprostowania do tego wniosku. Ale trzymajmy się porządku, dobrze? Tak, będzie pan miał głos po jeszcze dwóch wnioskach formalnych. Bardzo proszę, panie pośle. Dziś w wielu polskich domach gości strach i niepewność. Odpowiedzialny rząd dzisiaj powinien wyjść naprzeciw temu i dzisiaj przede wszystkim, panie premierze, nie podsycać tych niepokojów, tego strachu, wprowadzając niepewność, uspokajać sytuację. Dzisiaj polscy rodzice oczekują wiedzy, kiedy będzie lockdown i czy dzieci będą chodziły do szkoły, czy nie. Niech się pani uspokoi. Oczekują dzisiaj wiedzy, kiedy i jakie dziedziny będą działać. Polskie społeczeństwo oczekuje dzisiaj, jaka będzie hierarchia ważności celów podejmowanych przez władzę publiczną w Polsce. Nie oczekują, panie premierze, z całym szacunkiem, podsycania tej nienawiści, prowokowania do zachowań, które będą dalej prowadziły do wojny polskiej, wojny polsko-polskiej. Apelujemy do większości sejmowej, do polskiego rządu o łagodzenie nastrojów, o uspokajanie (Dzwonek) sytuacji, a nie o ich podsycanie. Dziękuję.

Wysoka Izbo! Wniosek formalny o przerwę i wprowadzenie do porządku informacji pana wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo.

Wszyscy powinniśmy odpowiadać za bezpieczeństwo. Myślę, że taka informacja od pana prezesa Kaczyńskiego, pana premiera - odpowiedzialnego za bezpieczeństwo - dałaby nam poczucie tego, że nie padają tu tylko słowa, ale że chodzi rzeczywiście o bezpieczeństwo. I apel do pana marszałka Terleckiego. Prosiłbym, żeby pan marszałek traktował równo Lewicę i opozycję, tak samo jak PiS. Chcę panu przypomnieć, że nie za pokrzykiwanie, tylko za blokadę mównicy sejmowej. Jeszcze przed panem pan poseł Janusz Korwin-Mikke z wnioskiem formalnym. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Popieram wniosek o przedstawienie nam sytuacji bezpieczeństwa i nie zgadzam się z Jarosławem Kaczyńskim, że Lewica działa dla małych, brudnych interesów. Działa dla zrobienia w Polsce rewolucji. Ci ludzie świadomie prowokują rewolucję.

Bo niestety w tej chwili sytuacja jest rewolucyjna. Przejęcie władzy przez Lewicę, rewolucyjną Lewicę.

Kobieta ma 300 razy większą szansę, że wpadnie pod samochód, idąc na protest, niż znajdzie się w sytuacji, w której urodzi kalekie dziecko. W trybie sprostowania. Odnoszę się do słów pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Prawda jest taka, że wyszedł podpalacz na mównicę i mówi: gasić pożar. Taka jest sytuacja dzisiaj w Polsce. To, co dzieje się na ulicach polskich miast, w Łodzi, Warszawie, Sieradzu, Zduńskiej Woli, Rzeszowie, to jest skutek pana działania. To, co obserwowaliśmy na sali sejmowej, to jest skutek pana działania. To jest skutek tego, że upolityczniliście Trybunał Konstytucyjny, że dzisiaj Trybunał Konstytucyjny jest na pilota, tak jak wszystkie inne instytucje państwa, takie jak prokuratura, telewizja. A ja jeszcze raz panu mówię, że my chcemy prawdy. Polacy dzisiaj oczekują prawdy o epidemii. Ukrywacie prawdę. Nie chcecie do niej dopuścić, bo się jej boicie, bo to jest wasz największy wróg. Największym wrogiem pana, panie premierze Kaczyński, jest prawda. Pan o tym doskonale wie. Taki jest po prostu fakt. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020, druk nr 713. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Wobec tego proszę państwa o przystąpienie do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Powracamy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce ustawy o spółdzielniach. Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały z druku nr 701. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 701, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Za - 409, przeciw - 1, wstrzymał się 1. Sejm podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce ustawy o spółdzielniach. Powracamy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 676-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Andrzeja Szlachtę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Pragnę przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych z druku nr 676-A o rządowym projekcie ustawy z druku nr 643. Na wczorajszym posiedzeniu Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła 20 poprawek. Po dyskusji, w wyniku głosowania, wszystkie poprawki zostały przez komisję odrzucone. Rekomenduję w imieniu Komisji Finansów Publicznych odrzucenie tych poprawek i przyjęcie projektu ustawy w całości. Dziękuję, panie pośle. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 676. Komisja przedstawia wniosek mniejszości oraz w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.

Komisja wnosi o ich odrzucenie. Ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość wniosku mniejszości oraz poprawek 2. i 12. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wymienionych poprawek, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. We wniosku mniejszości wnioskodawca proponuje zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 10., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 15., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 676, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Wzywam Konwent Seniorów do ciemnego saloniku.

Wznawiam obrady. Powracamy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 675-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Panie pośle, odbyła się właśnie przerwa, a pan może wnioskować o przerwę, więc w tej chwili nie ma to sensu.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pragnę przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych z druku nr 675-A w sprawie rządowego projektu ustawy z druku nr 642. Na wczorajszym posiedzeniu Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła w pierwszej kolejności wniosek o odrzucenie przedmiotowego projektu ustawy. Komisja wniosek zaopiniowała negatywnie. Komisja wnioskuje o odrzucenie tego wniosku przez Wysoką Izbę. Następnie komisja rozpatrzyła 35 poprawek.

W konkluzji komisja rekomenduje przyjęcie w całości przedmiotowego projektu ustawy. Bardzo dziękuję. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 675. Komisja przedstawia również wnioski mniejszości, a także w dodatkowym sprawozdaniu wniosek o odrzucenie projektu ustawy oraz poprawki.

Komisja wnosi o odrzucenie wniosku o odrzucenie projektu ustawy. Ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość pozostałych propozycji. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy oraz 1. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Tak, panie pośle, tylko pana wniosek o przerwę albo przerwanie obrad. Ale nie ma pan innej możliwości złożenia wniosku formalnego.

Zachowujecie się jak.

Proszę zająć miejsce. A oni mają? Nie, też nie mają.

Panie premierze, pytali o pana pod Sejmem. Idą po pana. Nie ma teraz wniosku formalnego. Ale pan mi chce dać głos po punkcie, a ja chciałbym Sejm przekonać przed punktem, żeby głosowali inaczej. Ale to nie jest wniosek formalny. A przerwa przed chwilą była. Proszę usiąść na miejscu.

Ja się nie boję. Jak ktoś ma czyste sumienie, to się nie boi.

Jasne, po tym głosowaniu, po tym punkcie dopuszczę pana do głosu.

Panie pośle, na podstawie art. 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję pana

Zobaczymy.

Ale nie ma takiej możliwości w czasie głosowań. Regulamin dopuszcza pytania.

A ja nie dopuszczam do pytań. Przeszkadza pan w głosowaniu. Zajmuje pan czas Sejmowi. Już pan złożył - o dopuszczenie pytań.

Ale to pan złożył wniosek. Niech pan składa.

Ta ustawa jest niezmiernie istotna. Państwo tą ustawą nakładacie nowe podatki na Polaków, którzy uzyskują dochody za granicą, oni nie mieszkają za granicą. Proszę sobie wyobrazić studenta, który np. studiuje w Wielkiej Brytanii i pracuje po to, żeby zarobić na studia. Proszę sobie wyobrazić Polaka, który np. przez 15 lat pracował na budowie w Irlandii, wrócił do Polski i uzyskuje emeryturę z Irlandii. Te dochody drugi raz w Polsce opodatkowujecie, drugi raz. Proszę sobie wyobrazić pracownika transgranicznego, który pracuje w kraju ościennym, a mieszka z rodziną w Polsce. Oni będą płacić podatki w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, w Norwegii i drugi raz jeszcze zapłacą podatek w Polsce.

Dziękuję.

W 1. poprawce wnioskodawcy proponują nowe brzmienie ustawy. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce nacisnąć przycisk? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił.

W 3. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują nie nadawać nowego brzmienia odpowiednim artykułom ustawy nowelizowanej.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Jego przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość 5. wniosku mniejszości. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Wniosek został odrzucony. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. wniosku mniejszości oraz tożsamej 2. poprawki, zechce nacisnąć

Sejm wniosek odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki? Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

Sejm poprawki przyjął.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem ww. poprawek?

Sejm wniosek odrzucił.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Sejm wniosek odrzucił.

Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił. Jego przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość 12. wniosku mniejszości oraz poprawek 11. i 12. Kto jest przeciw? się wstrzymał?

Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość 12. wniosku mniejszości oraz 12. poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11. poprawki?

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. poprawki?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 13. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 14. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 16. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 17. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosowało 441 posłów.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 18. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o odrzucenie poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 30. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 19. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił.

Przystępujemy do głosowania. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. W 20. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują zmianę terminu wejścia w życie ustawy. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 20. wniosku mniejszości? Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił. W 22. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują zmianę terminu wejścia w życie ustawy.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania.

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Tak jest, teraz właśnie jest czas na po jednym pytaniu każdego klubu. Bardzo proszę.

Wszyscy jesteście równie winni temu, że ci ludzie pracują za granicą, a nie pracują w Polsce. Cała klasa polityczna, która zarządza państwem przez ostatnie kilkadziesiąt lat, przyczyniła się do tego, że miliony Polaków pracują za granicą i niestety często muszą wyjechać - dla większości to nie był wybór na zasadzie fanaberii, dla większości to była jedyna szansa. Tak że wszyscy się do tego przyczyniliście, od lewa do tzw. prawa. I teraz macie szansę zagłosować przeciwko tej ustawie, macie szansę tych ludzi nie krzywdzić i macie szansę się na nich nie mścić za to, że postanowili wyjechać z Polski, żeby zarabiać normalne pieniądze. Dziękuję, panie pośle.

Przegłosowanie przez PiS tej ustawy to hańba.

Panie Kaczyński, jeśli wydał pan wszystkie pieniądze, to może pan swoją emeryturę dwa razy opodatkuje? Pan ma dochody jako poseł, ma pan dochody jako dietę, i ma pan jeszcze prawie 100 tys. zł emerytury rocznie, i płaci pan raz podatek. a Polak, który pracuje w Wielkiej Brytanii, będzie płacił dwa razy podatek. Dlaczego? Nie rozmawiacie z kobietami, nie rozmawiacie z rolnikami, nie rozmawiacie z ludźmi pracującymi za granicą, a potem się dziwicie, że oni tu wszyscy przychodzą i mają do was pretensje.

Panie pośle, proszę zająć miejsce.

Panie i Panowie Posłowie!

Dzisiaj zamiast od rządu Zjednoczonej Prawicy otrzymać pomocną dłoń, oni widzą gest Lichockiej, dostając podwójne opodatkowanie. Rząd ma 13 mld na Centralny Port Komunikacyjny - dzisiaj decyzja, o czym wasza telewizja informuje - a przedsiębiorcy będą gnębieni. Wymierzyliście już wyrok na rodzinne gospodarstwa rolne, teraz są przedsiębiorcy pracujący w spółkach komandytowych. Jest pytanie: Czy pomysłem Zjednoczonej Prawicy na walkę z kryzysem gospodarczym jest likwidacja przedsiębiorstw? Bardzo proszę. Wysoki Sejmie! Dzisiaj z jednej strony rząd mówi tak: trzeba chronić miejsca pracy, trzeba pomagać, trzeba walczyć o to, żeby przedsiębiorcy mogli funkcjonować - a z drugiej strony przedstawiacie projekt ustawy, który podnosi podatki, który opodatkowuje spółki komandytowe, który opodatkowuje osoby i Polaków, którzy pracują za granicą. Jaki jest w tym sens i jaka jest w tym logika? Mówicie oczywiście, że trzeba spółki komandytowe opodatkować, bo to kapitał zagraniczny.

Ale mamy teraz moment na pytania. W związku z czym mam jasne i klarowne pytanie do większości Prawa i Sprawiedliwości: Czy macie wyliczone, ile spółek komandytowych przez tę decyzję upadnie, ile miejsc pracy zostanie zlikwidowanych w Polsce, jeżeli tę ustawę dzisiaj przyjmiecie? Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę podsekretarza stanu w ministerstwie finansów pana ministra Jana Sarnowskiego. Bardzo proszę, panie ministrze.

Wysoka Izbo! Im dłużej słucham wypowiedzi posłów opozycji, tym bardziej mi się wydaje, że mówimy o dwóch całkowicie różnych projektach. Szanowni państwo, proponowana ustawa ma jeden bardzo konkretny cel. poprawę kondycji sektora firm małych i średnich w szczególnie trudnej sytuacji związanej z COVID-em. Przedsiębiorcy tracą i tracą nie tylko w wyniku związanych z epidemią ograniczeń, ale również w wyniku nowego zagrożenia, jakim jest niestabilność na rynku. Potrzeba trzech rzeczy, i to tych trzech rzeczy, które da im teraz ta ustawa. Po pierwsze, niskich podatków, takich, które pozwolą firmom na tworzenie finansowych poduszek bezpieczeństwa [[Oklaski]] i inwestowanie wtedy, kiedy jest to dla nich możliwe i korzystne. Stąd takie rozwiązania jak głosowany dzisiaj estoński CIT, poszerzenie dostępności ryczałtu. Oczywiście. Natomiast również obniżenie, poszerzenie możliwości zastosowania 9-procentowej stawki CIT-u dla dużej rzeszy przedsiębiorców. Po drugie, firmy potrzebują bezpieczeństwa, maksymalnej prostoty rozliczeń, tak żeby wykonywanie przez nie obowiązków związanych z podatkami zajmowało jak najmniej czasu i nie niosło ze sobą ryzyk. Pamiętajmy, im prostsze zasady rozliczenia podatku, tym niższe koszty jego obsługi.

warunków konkurencji. Chciałbym powtórzyć, że w trakcie spowolnienia gospodarczego, w trakcie wzmożonej rywalizacji między dużymi a małymi firmami należy zapewnić tym mniejszym podmiotom równe warunki konkurencji, a bardzo ważnym elementem przewagi konkurencyjnej dużych podmiotów są szerokie możliwości oszczędzania przez nie na podatkach, co jest skutkiem wypychania mniejszych firm przez większe z rynku. Chciałbym jeszcze raz mocno podkreślić, że prezentowany dzisiaj projekt, całość pakietu - i ten, nad którym państwo głosowali chwilę temu, i ten, nad którym głosować państwo będą za chwilę - to jest 7 mld zł w kieszeniach przedsiębiorców w przyszłym roku. Tylko w 1/4 koszt tego będzie pokryty przez zmiany uszczelniające podatki, przy czym uszczelnienia w ogromnej większości dotyczyć będą agresywnych optymalizacji związanych z wyprowadzaniem środków do rajów podatkowych. Na zmianach skorzysta 400 tys. firm, i to tych najmniejszych, dla których obniżka podatków stanowić będzie być albo nie być w trudnej walce o utrzymanie się na rynku. Jak najbardziej.

Nie dotyczy to tylko i wyłącznie 3% spółek komandytowych, które są własnością podmiotów zagranicznych.

Dotyczy to np. takich firm, których właścicielami są Polacy, które są zarejestrowane w rajach podatkowych, a w których Polacy są np. członkami zarządów. Szanowni Państwo! To, na czym nam zależy, to jest wyrównanie poziomu opodatkowania pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będącą partnerem spółki komandytowej w sytuacji, w której w obu tych spółkach za działalnością gospodarczą stoi tak naprawdę ta sama osoba. W takim schemacie spółka komandytowa kamufluje jedynie rzeczywistą działalność przedsiębiorcy, która w ogóle nie różni się od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to dokładnie to samo zjawisko, które koledzy z Platformy Obywatelskiej chcieli zlikwidować, uniemożliwić w roku 2013. Zrobiono to tylko w połowie wobec spółek komandytowo-akcyjnych mimo sprzeciwu Prawa i Sprawiedliwości oraz mimo sprzeciwu koalicjanta PSL-u. Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!

Zrobiło to już 12 państw Unii Europejskiej, na Zachodzie Belgia i Hiszpania, a w naszym regionie Litwa, Czechy, Węgry, Rumunia. Chcę bardzo mocno podkreślić, że objęcie CIT-em spółek komandytowych nie będzie oznaczało konieczności ich likwidacji, będą dalej służyć biznesowi do pozyskiwania kapitału, nie będą jedynie umożliwiać unikania opodatkowania. Mniejsze firmy nie odczują żadnej zmiany, CIT zapłacony przez spółkę będzie odliczany od podatku płaconego przez wspólników. Sytuacja komplementariusza się nie zmieni, bo dokona takiego odliczenia (Dzwonek), a komandytariusz skorzysta z kwoty wolnej od podatku.

Z kolei w przypadku spółek komandytowych, które są wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem jako narzędzie poszukiwania dodatkowego kapitału w spółce od podmiotów niepowiązanych, opodatkowanie spadnie z 19 na 17,29% u komplementariusza, również mniej podatku zapłaci komandytariusz tak długo, jak jego dochód nie przekroczy 156 tys. zł rocznie.

Szanowni państwo, rzeczywiście od roku 2008 r. obowiązują przepisy, które preferencyjnie traktują dochody osób, które mieszkają w Polsce, ale przez mniej niż 6 miesięcy w roku działają za granicą.

Co gorsza, ulga abolicyjna bardzo często służy nieuczciwym firmom, żeby w ogóle nie płacić podatków w Polsce.

Raz jeszcze chciałem państwu przypomnieć. że zmiany dotyczące ulgi abolicyjnej nie będą dotyczyć Polonii, nie będą dotyczyć 2,5 mln Polaków, którzy mieszkają w innych krajach Unii Europejskiej i na świecie. Będzie to dotyczyć tylko tych osób, które ponad 183 dni w roku mieszkają w Polsce i na krótszy okres niż pół roku wyjeżdżają za granicę. Takich osób są nie miliony, a 67 tys., przy czym zmiana w prawie, dzięki zastosowaniu kwoty wolnej od podatku, obejmie tylko 1/3 z nich, czyli niewiele ponad 20 tys. osób. Średnio więcej niż 10 tys. zł rocznie, a w 80% te dochody są przez nie osiągane w innych rajach podatkowych, czyli w Luksemburgu, na Cyprze i w Holandii. Podkreślam, studentów w ogóle to nie dotknie, ponieważ studenci objęci są PIT-em zero dla młodych już od zeszłego roku, na pewno państwo zdążyli to zauważyć.

Równamy do średniej europejskiej, nowego standardu wdrażanego w ogromnej większości państw Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z brzmieniu z druku nr 675, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo! Ale również otrzymaliśmy informację, że zajętych jest 1150 respiratorów. Na Mazowszu, szanowni państwo, jest wolnych 12 respiratorów. W Małopolsce jest wolnych 12 respiratorów. Nie wiemy, jakie są scenariusze i czy w najbliższych dniach nie będzie ogłoszony stan nadzwyczajny. Panie Premierze! Apeluję do pana, aby poprosił pan ministra Niedzielskiego, żeby złożył tu informację. Strategia, którą przedstawiliście, to jest pięć stron. Z niej nic kompletnie nie wynika. To nie był wniosek formalny, panie pośle. Słucham? Pan poseł Adam Szłapka, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Bardzo proszę na podstawie regulaminu o przerwę i informację marszałka Sejmu oraz premiera Morawieckiego o sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa. Z Sejmu zrobiliście twierdzę.

To są metody stosowane na Białorusi.

A pan nawołuje swoich zwolenników do wyjścia na ulicę. Pan nas nazywa przestępcami. To pan jest przestępcą. Ten okrzyk to był pana, panie pośle? Sprawdzimy.

Poddam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

A pan, panie pośle, po tylu latach mógłby się potrafić zachować na sali obrad. Właśnie widzę.

Dobra, panie pośle.

Za wnioskiem głosowało 210, przeciw - 234, 9 osób wstrzymało się od głosu. Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 23. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 712 i 713)

Wysoka Izbo! Do nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 Senat wniósł cztery poprawki. Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała poprawki. Rekomenduję Wysokiej Izbie odrzucenie trzech poprawek, a przyjęcie jednej. Dziękuję. Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. W punkcie porządku dziennego dotyczącym rozpatrywania poprawek Senatu głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu.

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki? Kto się wstrzymał?

Programy polityki zdrowotnej, zwiększyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2 mld zł. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 3. poprawce Senat proponuje utworzenie nowej rezerwy celowej: Środki na obsługę długu Skarbu Państwa, a także uzupełnienie środków na rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Powracamy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 670-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoki Sejmie! W dniu wczorajszym sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrzyła poprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W trakcie drugiego czytania zgłoszonych zostało 7 poprawek. Wszystkie poprawki mają charakter porządkowo-legislacyjny. Komisja Gospodarki i Rozwoju rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie tych poprawek. Dziękuję, panie pośle. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności.

Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z brzmieniu z druku nr 670, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 652-A.

Wysoka Izbo! Do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa w trakcie drugiego czytania złożono 15 poprawek. W dniu dzisiejszym Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyły te poprawki i rekomendują Wysokiej Izbie: poprawki 1., 2., 7. i od 9. do 15., głosowane łącznie, przyjąć, poprawki 3., 4., 5. i 8. odrzucić oraz przyjąć poprawkę 6. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 652. Komisje przedstawiają również poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.

Przystępujemy do głosowania.

Sejm poprawki odrzucił.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki? Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania.

Kto się wstrzymał?

Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 652, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Powracamy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 660-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Krzysztofa Szulowskiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Na posiedzeniu Sejmu w dniu wczorajszym zgłoszono trzy poprawki do projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, druki nr 512 i 660. W dniu dzisiejszym Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zebrała się w tej sprawie i rekomenduje przyjęcie każdej z tych poprawek. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki?

Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosowało 441 posłów. Sejm poprawkę przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki?

Za - 441, przeciw - 2, wstrzymało się 3. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 660, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 671-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Marka Asta o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo!

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 671. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm będzie głosować w pierwszej kolejności. W poprawkach od 1. do 4. wnioskodawcy proponują zmiany dotyczące zniesienia wymogu posiadania przez aplikanta aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej wyłącznie obywatelstwa polskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu druku nr 671, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 662. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 662? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty. Proszę pana posła Pawła Rychlika o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Dziś na posiedzeniu Komisja Zdrowia rozpatrywała rządowy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, druk nr 238. Komisja poprawkę 28. zaopiniowała pozytywnie, pozostałe - negatywnie. Komisja prosi Wysoką Izbę i rekomenduje przyjęcie całości projektu ustawy. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 663.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Kto się wstrzymał?

Za - 89, przeciw - 242, wstrzymało się 121 osób. Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2 poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał od głosu?

Za - 92, przeciw - 231, wstrzymało się 128 osób. Sejm poprawkę odrzucił.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Przystępujemy do głosowania.

Kto się wstrzymał?

Głosowało 450 posłów. Za - 208, przeciw - 242, nikt nie wstrzymał się od głosu. Sejm poprawki odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 4., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Za - 209, przeciw - 233, 12 posłów wstrzymało się od głosu. Sejm poprawkę odrzucił. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 5. i 7., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosowało 450 posłów. Za - 80, przeciw - 233, wstrzymało się 137 posłów. Sejm poprawki odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Sejm poprawkę odrzucił. Z poprawką tą łączy się poprawka 10. Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Za głosowało 161, przeciw - 234, 58 osób wstrzymało się od głosu. Sejm poprawkę odrzucił. Z poprawką tą łączy się poprawka 15. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 12. i 15., zechce nacisnąć przycisk.

Za - 205, przeciw - 243, nikt nie wstrzymał się od głosu. Sejm poprawki odrzucił. Z poprawką tą łączy się poprawka 16. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 13. i 16., zechce nacisnąć przycisk.

Za - 207, przeciw - 244, nikt nie wstrzymał się od głosu. Sejm poprawki odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 14., zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 17., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Za głosowało 205, przeciw - 242, wstrzymała się 1 osoba. Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Głosowało 449 posłów. Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 19., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 21., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 22., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 23., zechce nacisnąć przycisk. jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 24., zechce nacisnąć przycisk.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 25., zechce nacisnąć przycisk.

Za - 78, przeciw - 243, wstrzymało się 126 osób. Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 26., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 27., zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 28., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Za - 442, przeciw - 3, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Sejm poprawkę przyjął.

Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 30. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 29., zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 30., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Za głosowało 161, przeciw - 278, 10 osób wstrzymało się od głosu. Sejm poprawkę odrzucił.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 31., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 33., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Za - 167, przeciw - 278, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Sejm poprawkę odrzucił.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 36., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Za - 170, przeciw - 277, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 37., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Za - 170, przeciw - 276, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 38., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Za - 200, przeciw - 236, wstrzymało się 12 osób. Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 39., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem. Bardzo proszę. Panie i Panowie Posłowie!

To mogła być bardzo dobra ustawa, niestety jest tam kilka zapisów, które nas niepokoją.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 663, wraz z przyjętą poprawką, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zawodzie farmaceuty. Wysoki Sejmie! Czekają nas jeszcze głosowania zarówno proceduralne, jak i merytoryczne, więc informuję o tym. Grupa posłów przedłożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID. Zaraz do tego przejmiemy. To jest druk nr 717. Na posiedzeniu Konwentu Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec propozycji uzupełnienia porządku dziennego o pierwsze czytanie tego projektu. Jest to w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu punkt sporny porządku dziennego. Propozycję uzupełnienia porządku dziennego o ten punkt poddam pod głosowanie.

Wysoka Izbo! Wczoraj połączyła nas ponad podziałem politycznym ważna kwestia, wszyscy chcieliśmy pomóc pracownikom ochrony zdrowia, lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim bohaterkom i bohaterom, którzy stoją na pierwszej linii frontu walki z COVID-em. Dzisiaj, niespełna 12 godzin później Prawo i Sprawiedliwość chce tą ustawą okraść tych wszystkich, których wczoraj nagrodziliśmy za ich ciężką pracę. Ta ustawa to jest ustawa złodzieja, który chce po cichu odebrać pieniądze ludziom, którzy walczą o nasze zdrowie. Premier Morawiecki i minister Niedzielski w tamtym tygodniu z tej mównicy mówili: będziemy pomagali tym ludziom, będziemy stali po ich stronie. Pytam się: Po jakiej stronie stoicie? Panie Premierze! Mówię do pana premiera Kaczyńskiego. Czy bezpieczeństwo obywatela to nie jest też bezpieczeństwo walki o to, żeby ci ludzie więcej zarabiali? Czy nie chodzi o to, żebyśmy dawali im pieniądze, mając świadomość, że oni swoją ciężką pracą się poświęcają? Tu nie chodzi o to, żebyśmy się przekładali: czy prawica, czy lewica. Tu chodzi o uczciwość. Szanowni Państwo z PiS! Stańcie po stronie ludzi, którzy walczą o nasze zdrowie. Oni na to zasługują. Dziękuję bardzo.

Ja już pomijam ten język, którego lepiej by nie stosować w tej Izbie. Ale myśmy się już do tego przyzwyczaili.

Ale to jest tylko kwestia poboczna. Wzywałbym do tego, żeby wrócić chociaż do obyczajów tej lewicy, której tutaj już nie ma. Bo chociaż były złe, to jednak nieporównanie lepsze niż wasze. To sprawa pierwsza. Ale sprawa druga. Państwo, a właściwie wasze kluby parlamentarne, wasi senatorowie, marszałek Senatu przeprowadzili w Izbie wyższej zmianę (Dzwonek), która w gruncie rzeczy sprowadza się do dwóch punktów. Po pierwsze, do tego, że ten, kto przez telefon udziela porad i nawet nie widuje się z chorymi, i ten, który ryzykuje, walcząc bezpośrednio z COVID-em, mają być potraktowani tak samo. A po drugie, to prowadzi do dodatkowych 40 mld, to znaczy do zniszczenia Narodowego Funduszu Zdrowia. i do zniszczenia całych finansów publicznych. Być może Janusz Korwin-Mikke miał rację, że też ideologicznych, ale przede wszystkim tych małych.

Panie marszałku, prosiłbym o taki sam przydział czasu, jak miał pan prezes Kaczyński, bo jesteśmy w tym Sejmie równi. Pozbawiliście znaczną część lekarzy dodatków i Senat te dodatki przywrócił. I ta poprawka jest bardzo słuszna, ale mam złą wiadomość dla PiS i bardzo dobrą wiadomość dla lekarzy, bo chcieliście zabrać dodatki za pracę na oddziałach zakaźnych, ale wydaje się, że to będzie niemożliwe.

Chciałbym państwa poinformować, poinformować Wysoką Izbę, że taka ustawa nie weszła w życie. Nie można zmienić ustawy, która nie weszła w życie. Ta ustawa nie wyszła z Sejmu, nie dotarła do prezydenta, prezydent jej nie podpisał. W związku z tym nie można jej zmienić. Dziękuję, panie pośle. Wyczerpał pan czas. Macie państwo większość w tej Izbie, więc chociaż ustawy mogłyby być przegłosowywane większością - prawdziwe ustawy. A państwo proponują dzisiaj państwo bez żadnego trybu. Pan poseł Michał Szczerba, klub Koalicji, z wnioskiem formalnym.

Chciałbym na chwilę te wszystkie emocje tej Izby wyciszyć, ponieważ chciałbym przypomnieć o ważnej rocznicy. Dzisiaj, Wysoka Izbo, jest 7. rocznica śmierci pierwszego niekomunistycznego premiera Tadeusza Mazowieckiego. Tadeusz Mazowiecki był wieloletnim posłem, ale był pierwszym niekomunistycznym premierem. Był człowiekiem dialogu, człowiekiem mądrości, człowiekiem kompromisu.

Pan poseł Krzysztof Paszyk z wnioskiem formalnym.

Wysoka Izbo! Na początek, panie prezesie, wezmę trochę w obronę koleżanki i kolegów z Lewicy, bo przykro to powiedzieć, ale pan też ma swój udział w tym... ...komuna. Natomiast, panie prezesie, jako lider większości sejmowej, większości zasiadającej na tej sali, ponosi pan też odpowiedzialność za to, jak Polacy będą postrzegać jakość naszej pracy. Dzisiaj już mleko się rozlało. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni wczoraj doskonale zorientowali się, że przyjęto jakieś rozwiązanie prawne.

Dziękuję bardzo. Zwracam uwagę, że to nie był wniosek formalny. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowanie to nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Przyjęcie propozycji uzupełnienia porządku dziennego oznaczać będzie, że Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu Sejmu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk nr 717), zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosowało 441 posłów. Sejm propozycję przyjął. Proponuję, aby Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła w dyskusji nad dodanym punktem porządku dziennego. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Poddam go wobec tego pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem propozycji wysłuchania 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 24. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk nr 717) Proszę pana posła Jacka Żalka o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Projekt tej nowelizacji jest bardzo poważny. Poważny dlatego, że chcieliśmy docenić pracę tych, którzy ratują życie i zdrowie naszych rodaków. którzy nie mają tyle szczęścia, żeby ocalić swoje zdrowie, a czasami życie, przed tą epidemią. Dlatego potrzebujemy docenienia pracy lekarzy i tych wszystkich, którzy na pierwszej linii w służbie zdrowia niosą pomoc naszym rodakom. Sytuacja, w której Wysoka Izba przyznaje wszystkim dodatek, niezależnie od tego, czy się angażują, tylko dlatego, że są pracownikami służby zdrowia, co wyklucza możliwość różnicowania i docenienia pracy tych, którzy naprawdę się poświęcają, jest niestety kpiną.

pracują, angażują się, narażają się, a nie wszystkim, bo to wyklucza możliwość wyróżnienia tych, którzy są na pierwszej linii frontu. Jeżeli to uzasadnia awanturę w parlamencie, to w takim razie jakie można inne racje przedstawić? Czy zależy nam na tym, żeby środki, którymi dysponujemy, jak najlepiej, jak najcelniej, najtrafniej przeznaczyć na potrzeby tych, którzy niosą pomoc naszym chorym, czy też żeby je jak najszybciej roztrwonić? To pytanie, oczywiście, jest pytaniem retorycznym. Widzę, że nie ma atmosfery w ławach opozycyjnych do prowadzenia debaty.

Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu pozytywnie odnoszące się do propozycji zaprezentowanych w poselskim projekcie ustawy z druku nr 717 i jednocześnie wnoszę o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania. Bardzo dziękuję. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska pan poseł Borys Budka. Panie Marszałku! Nie potraficie przyjąć dobrych rozwiązań i po raz kolejny dzielicie Polaków, tym razem lekarzy. Kochani, nie ma żadnej różnicy, czy ktoś pracuje w walce z COVID-em w takim, a nie innym szpitalu. Kłamaliście rano, kłamiecie w południe i potraficie kłamać wieczorem. Jesteście bandą hipokrytów, która kolejny raz chce okradać Polaków. Gdzie byliście, kiedy rozdawaliście miliony Rydzykowi? Gdzie byliście, kiedy wasz kolega zamawiał bez przetargów respiratory? Gdzie byliście wtedy? Okradaliście Polaków, a dzisiaj chcecie okraść polskich lekarzy. Wczoraj przyjmujecie ustawę, dzięki której i dzięki opozycji daliśmy środki wszystkim według tego, że walczą z COVID-em, ale wy musicie zabrać, bo wy nie potraficie przyjąć jednego prawa, które jest sprawiedliwe dla wszystkich. Bo wy się czujecie jak ci władcy, którzy mają taką moc, żeby dawać, ale tylko wybranym. W zamierzchłych czasach może tak, ale pan swoją działalnością udowadnia, że ten doktorat powinien być panu dawno odebrany, bo nikt nigdy nie podeptał polskiej konstytucji tyle razy, ile pan i pana koledzy.

W imieniu klubu Lewicy pan poseł Jan Szopiński. Bardzo proszę. W tej chwili cały medyczny personel, który zmaga się z przeciążeniem i niewydolnością systemu, który walczy z czasem, presją, brakiem spójnej i jasnej strategii rządu, ale też przecież z prawem i własnymi słabościami, odpornością na stres i wielką odpowiedzialnością, potrzebuje przede wszystkim wsparcia, potrzebuje testów, szacunku, motywacji, pomocy w budowaniu społecznego zaufania, ale też potrzebuje wsparcia finansowego. A wy co robicie? To zawsze najlepiej wam wychodzi i w sposób absolutnie haniebny chcecie zmienić uchwalone przez Sejm wczoraj przepisy. Robicie wrzutkę, nowelizację do nieistniejącego prawa. Nie jesteście w stanie zapanować nad chaosem, bo nigdy nie zapewniliście obywatelom bezpieczeństwa i przemyślanej konsekwentnej strategii walki z pandemią. Dziś zbieramy żniwo waszych zaniechań i skrajnej nieodpowiedzialności. Chaos w służbie zdrowia pogłębia się coraz bardziej, z godziny na godzinę. Strach obywateli jest coraz większy. Gdyby nie ludzie, którzy walczą na pierwszej linii frontu z COVID-em, lekarze, ratownicy, pielęgniarki, diagności, laboranci, już dawno załamałby się system zdrowia.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polska służba zdrowia marzyła o tej ustawie, która dawała środki finansowe zarówno lekarzom kierowanym przez wojewodów do jednostek służby zdrowia, jak i tym, którzy w tych jednostkach zdrowia są zatrudnieni. To była szansa i okazja do tego, aby z jednej strony te środki trafiły do lekarzy, z drugiej strony trafiły do pielęgniarek, do osób z personelu medycznego średniego, których ogromnie wiele jest w takim szpitalu, bo są to kucharki, są to salowe, dodatkowo jeszcze jest personel, który decyduje o badaniach w szpitalach. Oni wszyscy mieli otrzymać stosowne dodatki, mieli otrzymać te dodatki niezależnie od tego, jaki jest stopień ich zatrudnienia. Natomiast chciałbym zapytać: Co stało się dzisiaj od godz. 24 do dzisiejszego dnia? Co znaczy owo słowo „konwalidacja” Chciałbym te pytania zadać panu, panie prezesie. Czyżby znaczyło to, że teraz oni są przeciwko polskiej służbie zdrowia? Dodatkowo, szanowny panie prezesie, gdybym ja miał - w zestawie tych, którzy popełniają taką pomyłkę - jednego wicepremiera, jednego ministra, jednego wiceministra, tobym się zastanowił, czy ci ludzie powinni pełnić te funkcje.

Jest na tej sali jedna poseł, znana bynajmniej nie z gestów parlamentarnych. A teraz czytam w uzasadnieniu tego projektu, że się podpisuje: nie dajmy pieniędzy służbie zdrowia. Chciałbym zapytać: Kiedy ona jest po prostu poważna? Natomiast, wie pan, panie prezesie, jestem z Kujaw i Pomorza.

Takich pomyłek nie powinno być. Chciałbym. na ręce pana marszałka [[Dzwonek]] złożyć wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, bo tego oczekuje polska służba zdrowia. W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego pan poseł Władysław Kosiniak-Kamysz. Po pierwsze, panie marszałku, w imieniu klubu Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Następnym razem marszałek Zgorzelski pana będzie przedstawiał jako przedstawiciela Porozumienia. To jest pierwsza kwestia. Po pierwsze, kpicie z parlamentaryzmu i wczorajszej decyzji Sejmu. Również waszej, bo za nią głosowaliście. Nie kpijcie z nich. Obiecaliście im, bo to mówił minister Niedzielski na moje pytanie na ostatnim posiedzeniu Sejmu, czy premie będą dla wszystkich. Nie tylko dla tych skierowanych przez wojewodę, nie tylko dla tych, którzy pójdą do Szpitala Narodowego. Dla wszystkich, którzy będą leczyć chorych na COVID-19. I ta premia im się należy nie od dziś, nie od wczoraj, tylko od marca 2020 r., kiedy rozpoczęli walkę na pierwszej linii frontu. Salowe, ratownicy medyczni, diagności, fizjoterapeuci, pielęgniarki i lekarze. To są współcześni bohaterowie. W nocy głosujecie: tak, dajmy im więcej pieniędzy. Wynagrodźmy to staranie, które oni oddają każdego dnia. To ryzyko dla siebie, dla swojej rodziny. Również wynagrodźmy tych, którzy poświęcili swoje zdrowie, bo zachorowali na COVID-19, bo leczyli, bo ratowali zdrowie i życie. Ale tu nie ma szacunku dla zdrowia i życia. Jest utrata kontroli nad państwem. Utraciliście kontrolę nad epidemią, utraciliście kontrolę nad państwem, ale - co więcej - utraciliście kontrolę nad większością. Bo wczoraj większość przegłosowała to. Im się to po prostu należy. Tak jak kiedyś wasza premier mówiła, że i wam się należały premie w ministerstwach. To oddajcie te premie, które dała Emilewicz, odchodząc, i dajcie je na lekarzy, na pielęgniarki, na ratowników. Jeżeli komuś się dzisiaj w Polsce coś należy, to na pewno należy się szacunek, wdzięczność i godne wynagrodzenie dla bohaterów, którzy ratują nasze życie i zdrowie. Nie możecie tego zrozumieć.

Głosowaliście, bo może mieliście przebłysk przyzwoitości. Dzisiaj trzeba wnosić o odrzucenie. O odrzucenie tej ustawy w całości, bo niestety nie potraficie jednego. Nie potraficie jednego: zrozumieć, że trzeba docenić tych, którzy poświęcają swoje życie i zdrowie. Wy nie jesteście w stanie tego zrozumieć, bo dzisiaj wnosicie cyniczną ustawę, która na pierwszym miejscu stawia tylko i wyłącznie wasz interes. Dzisiaj ci pracownicy utrzymują sprawność ochrony zdrowia. Odrzucić to w całości.

Wysoka Izbo! Uzasadnienie do tej ustawy napisanej jakoś tak kilkanaście minut temu: celem projektu ustawy jest konwalidacja błędu, który miał miejsce podczas rozpatrywania w Sejmie poprawek Senatu do bla, bla, bla. Wystarczyło napisać trzy zdania. Szanowni lekarze, głosujcie na Konfederację i Korwina-Mikke. Oni obniżą wam podatki i będziecie wreszcie więcej zarabiać, bo my wam tego nie załatwimy. Szanowni Państwo! Po prostu spieprzyliście, no. Tyle. Zagłosowaliście źle. Po prostu staliście i był sztab kryzysowy. Co się dzieje? Trzeba było szybciutko zareagować. Nie zareagowaliście, nie zareagowaliście na to niestety. i dzisiaj urządzacie tę szopkę z nową ustawą napisaną w 5 minut, naprawdę wyglądającą żałośnie. Przepchniecie to oczywiście, no jasne, że to przepchniecie, bo macie większość w tej Izbie. Ale wiedzcie, że to wygląda obrzydliwie. I dzisiaj, podczas tych protestów, które tam są na zewnątrz, z którymi ja się oczywiście nie zgadzam. Ja się troszkę boję, że mogą się tam przyłączyć lekarze po tej decyzji, którą zaraz podejmiecie. Wyznaczam czas pytania na 1 minutę.

Bo chcecie państwo głosować nad ustawą, w której są trzy kropki.

A jak ktoś tam pisze parę gwiazdek, które ludzie krzyczą na ulicach, to też zagłosujecie? Też wam się to będzie podobało? Mówiono o przyzwoitej legislacji. Tu nie ma ani przyzwoitej legislacji, ani zwykłej przyzwoitości. Nic nie powiedział, bo o tym nie da się nic powiedzieć. To jest zwykły bubel i bzdura. Powinniście się wstydzić, że w ogóle coś takiego przynosicie do Wysokiej Izby. Pan poseł Jarosław Rzepa, klub PSL. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Padły tutaj słowa, że powinniście się wstydzić. Pani poseł, moja żona pracuje w szpitalu COVID-owym na bloku operacyjnym i wiem, co robi każdego dnia. Wiecie, co było na początku? Nie chcieliście ich nawet wymazywać. żeby mogli mieć testy.

Mówicie, że dla nich nie ma pieniędzy. Słuchajcie, zrobiliście z tej Izby, nie wiem, cyrk. Szanowni państwo, niezakończony proces legislacyjny, a my chcemy to zmieniać. To jest Sejm? Tym ludziom, którzy od marca pracują, naprawdę się to należy. Pani poseł Krystyna Sibińska, klub Koalicja Obywatelska. Dostaję takie informacje z województwa lubuskiego: szpital w Drezdenku - nie ma sprzętu, nie ma respiratorów, nie ma jak leczyć, a wojewoda zrobił ten szpital szpitalem COVID-owym. W szpitalu w Gorzowie pielęgniarki są sekretarkami i osobami, które robią wymazy, bo brakuje ludzi, brakuje zaopatrzenia. Jak mamy im to wynagrodzić?

Trzeba docenić tych, którzy ciężko pracują. Ciężko pracują dlatego, że muszą to robić, bo mają poczucie misji, chcą to robić, a wy chcecie znowu dzielić. Dzielić na tych, których wyśle wojewoda, bo to będzie swój. A ci, którzy teraz ciężko pracują, nie są swoi i im się nie należy. Nie minął tydzień, a większość sejmowa polskiego parlamentu napluła w twarz kobietom, napluła dzisiaj w twarz przedsiębiorcom, którzy tworzą spółki komandytowe, i jeszcze w tym samym tygodniu napluła w twarz lekarzom i służbom medycznym. Drodzy Państwo ze Zjednoczonej Prawicy! Naprawdę ogarnijcie się, bo w innym przypadku taczki pod Sejmem za chwilę będą na was czekać. Ogarnijcie się, bo straciliście podstawowe zdolności kontroli nad tym, co się dzieje w państwie. Pani poseł Agnieszka Pomaska, klub Koalicji Obywatelskiej. Wysoka Izbo! Najpierw chciałam się zwrócić do wnioskodawców, bo widzę, że nie są zbyt aktywni w tej debacie, wstydzą się albo się boją. Być może pan poseł Macierewicz chciałby nam coś ciekawego powiedzieć. Taki aktywny był wczoraj i dzisiaj, a teraz widzę, że w sejmowych ławach przysypia. Być może w błąd wprowadziła go telewizja, tzw. telewizja publiczna za 2 mld zł. Chcę przypomnieć, że w Wysokiej Izbie leży projekt przeznaczenia 2 mld zł zamiast na kłamliwą telewizję na służbę zdrowia. Czy wolą, żeby leczyli ich tacy ludzie jak wy, którzy zmarnowali 70 mln na pseudowybory, którzy zmarnowali pieniądze na lipne respiratory, czy chcą, żeby ich leczyli bohaterowie: lekarze, pielęgniarki, przedstawiciele służby zdrowia?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Za afery respiratorowe, maseczkowe, testowe i z przyłbicami daliście swoim w Ministerstwie Zdrowia po 30 tys. premii. 30 tys. Nie urzędnikom tylko swoim. Tu medyków chcecie dzielić na lepszych i gorszych. Apeluję do was: Wycofajcie się z tego, bo jutro do protestujących dołączą medycy. Jeszcze jedno, korzystając z okazji. Nie ma pana wicepremiera Kaczyńskiego, ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Do czasu. Wycofajcie się. Proszę, pan poseł Jakub Rutnicki, klub Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Dzisiaj ponad 18 tys. zachorowań, ponad 236 zgonów. Wasz minister zdrowia, Szumowski, zdezerterował. A jaką macie propozycję dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych? To są ludzie, którzy zasługują na te pieniądze. A wy co robicie w tym momencie? Próbujecie jeszcze ich dzielić. To jest skandal. To jest hańba, bo za chwilę naprawdę nie będzie miał kto leczyć Polaków. Takimi decyzjami rujnujecie tak naprawdę służbę zdrowia, która jest absolutnie na skraju przepaści. Pani poseł Katarzyna Lubnauer, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie i Panowie Posłowie! 18 820 nowych zachorowań, 236 nowych śmierci to bilans dzisiejszego dnia. Ale wy już w tym piekle dawno powinniście być.

Powinniście być w piekle za to, że lato przespaliście, zajmowaliście się sami sobą, wyborami, wszystkim tym, co dotyczyło rekonstrukcji rządu. Tylko że ja bym na waszym miejscu przemyślała to i każdy z osobna niech się zastanowi, bo za moment być może życie jego lub jego rodziny będzie zależało od tych, których teraz chcecie okraść. Bo to, co robicie, to tą ustawą chcecie okraść lekarzy. Dlatego zagłosujcie za wnioskiem o odrzucenie tej ustawy w pierwszym czytaniu, który złożyliśmy, bo być może uratujecie życie kogoś z waszej rodziny.

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Premierze Kaczyński!

Po drugie, wszyscy pamiętamy obrazki z telewizji - sanitariusze cały dzień w kombinezonach, cały dzień bez posiłków, cały dzień opiekują się chorymi na COVID, cały dzień lekarze na dyżurach, 15, 20 dyżurów w ciągu miesiąca lekarzy na oddziałach zakaźnych. Państwo wczoraj daliście im pieniądze, powiedzieliście, że zasługują, a dzisiaj mówicie: nie, odbieramy wam to, czego jeszcze nie daliśmy. A telewizji dawaliście państwo każdego roku 2 mld zł. Bardzo dziękuję.

Panie premierze Kaczyński, dzisiaj my pytamy: Czy zna pan przysłowie: kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera? Pani poseł Ewa Kołodziej, klub Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Jeszcze nie tak dawno w kontekście młodych lekarzy z ust polityków PiS padały haniebne słowa: niech jadą. A w rządowej telewizji nagminnie oczerniano ich i mówiono o kanapkach z kawiorem i luksusach, w których rzekomo się pławią. Przypomnę: w mediach rządowych, na które przeznaczyliście z początkiem tego roku 2 mld zł. Dlaczego o tym mówię? Dlatego że szacowane koszty wejścia w życie dzisiaj po raz drugi proponowanej ustawy w kontekście podwyżek dla medyków to zaledwie 9 mln zł. To prawie 8 razy mniej niż majowe wybory Sasina, które się nie odbyły, to ponad 200 razy mniej, niż przeznaczacie rok do roku na propagandę w swoich mediach publicznych. Z uporem maniaka zatem będę pytać: Po czyjej stronie stanie rząd PiS-u, czy po stronie Polaków i ich zdrowia, czy po stronie Jacka Kurskiego? Proszę zatem odpowiedzieć obywatelom na najważniejsze pytania: Czy rząd w tak dramatycznej sytuacji pandemicznej zdobędzie się na odwagę i pieniądze. Dziękuję pani bardzo. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Zamykam dyskusję. W dyskusji zgłoszono wnioski: - o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, - o przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania. Do głosowania nad tymi wnioskami przystąpimy za chwilę.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 717, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Wniosek został odrzucony. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za niezwłocznym przystąpieniem do drugiego czytania projektu ustawy, zawartego w druku nr 717, zechce nacisnąć

Nie jest pan spokojny, znowu pan przeszkadza.

Tylko wy. Chodzicie, mówicie, ile macie głosów, ile wam brakuje.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. W związku z decyzją Sejmu przystępujemy do drugiego czytania. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w drugim czytaniu projektu? Tak, mamy zgłoszenia. Bardzo proszę.

Rozumiem, że sprzeciwu już nie słyszę. Pan poseł Michał Woś, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Niestety ta debata przerodziła się w jakąś szopkę i trzeba tak to nazwać - szopkę, którą urządziła opozycja.

Dlatego, że wystarczą dwie liczby: jedna - 77 mld. Już wielokrotnie przy każdej debacie o służbie zdrowia o tym mówimy, ale znowu chyba trzeba to powtórzyć.

Drodzy Państwo! Ta ustawa jest właśnie o wsparciu tych bohaterów, którzy są na pierwszej linii frontu, tych, którzy walczą z COVID-em, bezpośrednio walczą z COVID-em. I państwo zamiast wspierać, solidarnie wspierać dobro wspólne, wspierać też pewne ułożenie budżetowe, cynicznie wykorzystują ten moment. Osobiście to odbieram także jako osoba, która właśnie tym ludziom serdecznie dziękuje. Szanowni Państwo! Nie bądźcie cyniczni, bo walka z pandemią jest naprawdę czymś, z czym rząd Zjednoczonej Prawicy sobie radzi i poradzi, daj Panie Boże. Składam wniosek o niezwłoczne przejście w wyniku tych wszystkich emocji i manipulacji do trzeciego czytania. Bardzo dziękuję.

Dodatek nie tylko dla wybranych, dodatek nie tylko dla niektórych, dodatek nie tylko dla wyróżnionych, bo wszystkim tym, którzy walczą na pierwszej linii frontu z COVID-em w różnych szpitalach i placówkach, należy się 100% dodatkowego wynagrodzenia. Nie ma naszej zgody na podziały.